Otwieram posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Grzegorza Pudę, Waldemara Budę, Monikę Wielichowską i Krzysztofa Truskolaskiego. W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Grzegorz Puda i Waldemar Buda. Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Grzegorz Puda i Monika Wielichowska.

Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Żegnamy dziś naszego kolegę, przyjaciela - Pawła Adamowicza, człowieka, którego znaliśmy od zawsze.

Był bardzo odważny. Był człowiekiem odważnym, nie bał się walki, ale swoje życie poświęcił ukochanemu miastu Gdańskowi. On jako pierwszy z nas zaangażował się w samorząd, w lokalną władzę i zrobił to w wielki sposób, w wielkim stylu. Pawła zabiła nienawiść. Nienawiść obłąkana, nienawiść dobrze zorganizowana, nienawiść przeciwko człowiekowi, który razem z tysiącami gdańszczan budował swoje wielkie, wolne, dumne miasto. Ale także nienawiść przeciwko człowiekowi, który razem z milionami Polaków tak mocno angażował się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Zanim to światło do nieba dotarło, dotarła tam także jego dusza. Wtedy powiedział: To jest cudowny czas, czas dzielenia się dobrem. Chcę ci teraz, Pawle, obiecać w imieniu przyjaciół, koleżanek, kolegów z Platformy Obywatelskiej, nas wszystkich, że będziemy o tym pamiętać, że ta nienawiść, która odebrała ci życie, nie zniszczy tego wszystkiego, co zbudowałeś, nie zniszczy miłości do wolnej Polski, nie zniszczy twojego Gdańska i nie zniszczy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - tych wszystkich rzeczy, którym poświęciłeś swoje życie i za które swoje życie oddałeś.

Dziękuję panu posłowi. Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktów w brzmieniu:

Grupa posłów przedłożyła wniosek w sprawie wyboru sędziego Trybunału Stanu, druk nr 3115. Opinia komisji to druk nr 3125. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tej sprawy. Komisja Finansów Publicznych przedłożyła dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, druk nr 3021-A. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący trzecie czytanie tego projektu ustawy. Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3116. W związku z tym, na podstawie art. 95b regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu ustawy. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projektach ustaw: - o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Są to odpowiednio druki nr 3122 i 3131. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę rozumiał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projektach ustaw: - o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej. Są to druki nr 3000, 3126 i 3121.

Rada Ministrów przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3045. Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec propozycji uzupełnienia porządku dziennego o pierwsze czytanie tego projektu. Jest to, w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu, punkt sporny porządku dziennego. Propozycję uzupełnienia porządku dziennego o ten punkt poddam pod głosowanie. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3045, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm propozycję przyjął. Grupa posłów przedłożyła projekt ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, druk nr 3114. Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec propozycji uzupełnienia porządku dziennego o pierwsze czytanie tego projektu.

Kto z państwa jest za uzupełnieniem porządku dziennego o ten punkt, czyli o pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm propozycję przyjął. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół w dyskusjach nad punktami porządku dziennego. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę rozumiał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Informuję, że Konwent Seniorów jednomyślnie zaopiniował propozycję rozpatrzenia na bieżącym posiedzeniu informacji w sprawie pogarszającej się sytuacji w systemie opieki zdrowotnej, o której przedstawienie wnosił Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów. Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Informacja w tej sprawie, a także wykaz ustaw, które Senat przyjął bez poprawek, dostępne są w Systemie Informacyjnym Sejmu. Proszę pana posła sekretarza o odczytanie komunikatów.

Proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Panie Premierze! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! 14 grudnia 2018 r. na posiedzeniu plenarnym odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019. Podczas debaty zgłoszono wniosek o odrzucenie rządowego projektu ustawy budżetowej, jedną poprawkę do części tekstowej i 109 poprawek do załączników projektu ustawy budżetowej. W dniu wczorajszym Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła wniosek o odrzucenie projektu ustawy, 109 poprawek i poprawkę do części tekstowej.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił.

Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 17. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem 28. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z państwa jest za przyjęciem 34. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z państwa jest za przyjęciem 37. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z państwa jest za przyjęciem 38. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto się wstrzymał?

Kto z państwa jest za przyjęciem 121. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z państwa jest za przyjęciem 126. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem 128. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 130. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 130. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z państwa jest za przyjęciem 131. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem 136. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 141. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Głosujemy. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 146. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 146. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Głosujemy. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 148. wniosek mniejszości. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z państwa jest za przyjęciem 149. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z państwa jest za przyjęciem 152. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 156. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 156. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 157. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 157. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 158. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 159. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 159. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy.

Sejm wniosek odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Rozpatrujemy 164. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 164. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 165. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 165. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 31., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 166. wniosek mniejszości. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 167. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 167. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 168. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 168. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 33., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej odrzucenie.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 175. wniosek mniejszości.

Rozpatrujemy 177. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 177. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 178. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 178. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 179. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 179. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 180. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 180. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem 181. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 182. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 182. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 183. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 183. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 184. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 184. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Rozpatrujemy 47. poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem 48. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 49., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy 185. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 185. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 186. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 186. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 187. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 187. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 188. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 188. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 189. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 190. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 190. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 192. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 192. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 193. wniosek mniejszości. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 194. wniosek mniejszości. Głosujemy. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 195. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 50. poprawkę.

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 50., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 196. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 197. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 198. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 198. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Rozpatrujemy 199. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy poprawkę 52. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 52., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 414 posłów. Sejm wniosek odrzucił.

Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 202. wniosek mniejszości. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 203. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 203. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 204. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 204. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 205. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 205. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 206. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 206. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 207. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 207. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 208. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 208. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 209. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 209. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 210. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 210. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 211. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 211. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 212. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 213. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 214. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 215. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 215. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił.

Rozpatrujemy 54. poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 54., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Rozpatrujemy poprawkę 55. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 55., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Rozpatrujemy 56. poprawkę. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 216. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 216. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 218. wniosek mniejszości.

Kto z państwa jest za przyjęciem 219. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił.

Przechodzimy do rozpatrzenia 57. poprawki. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 57., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy 220. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 220. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy poprawkę 58. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 58., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Rozpatrujemy 59. poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z państwa jest za przyjęciem 59. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Rozpatrujemy poprawkę 60. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 60., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Rozpatrujemy 62. poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Rozpatrujemy 63. poprawkę. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy poprawkę 64. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 65. poprawkę. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 65., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy 66. wniosek mniejszości. Przepraszam, rozpatrujemy 66. poprawkę. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 66., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 67. poprawkę. Komisja wnosi o jej odrzucenie.

odrzucił.

Głosujemy. Kto z państwa jest za jego przyjęciem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Rozpatrujemy 238. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 238.

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 239. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Głosowało 410 posłów. Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 240. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za jego przyjęciem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z państwa jest za jego przyjęciem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 243. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 244. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 245. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 246. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 72. poprawkę. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy poprawkę 73. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy 74. poprawkę. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 74., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy poprawkę 75. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem 75. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy poprawkę 76. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 76., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy 77. poprawkę. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 77., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z państwa jest za jego przyjęciem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 248. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za jego przyjęciem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 249. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 78. poprawkę. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem tej poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy 250. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy poprawkę 79. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 79., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy poprawkę 80. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy 251. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 252. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 253. wniosek mniejszości.

Rozpatrujemy 254. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 254. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Rozpatrujemy 255. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Rozpatrujemy 256. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Rozpatrujemy 257. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 258. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 82. poprawkę. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 82., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy poprawkę 83. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 83., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy 84. poprawkę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy poprawkę 85. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 85., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy poprawkę 86. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 86., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 260. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 261. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 87. poprawkę. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 87. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 88., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 89., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy poprawkę 90. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 90., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy 262. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 262. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy 263. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 265. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za jego przyjęciem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił.

Wznawiam obrady. Proszę zająć miejsca.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 266. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 267. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 267. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 268. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 269. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 270. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 270. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 271. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 272. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 273. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 274. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 275. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 277. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 278. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 279. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 280. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 280. wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 281. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 282. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Rozpatrujemy 284. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem 287. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Rozpatrujemy 288. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 288. wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 289. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 292. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 293. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 294. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 295. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 296. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Rozpatrujemy 297. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 97. poprawkę. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 97., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy 298. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 299. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 300. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 300. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Głosujemy. Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 302. wniosek mniejszości. Kto się wstrzymał?

Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 304. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem 304. wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 305. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 307. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 308. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 309. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za jego przyjęciem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 310. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 311. wniosek mniejszości. Kto się wstrzymał?

Poprawki. Rozpatrujemy 98. poprawkę. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 98., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy 312. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za jego przyjęciem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 313. wniosek mniejszości. Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 314. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 315. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 316. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za jego przyjęciem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 317. wniosek mniejszości.

Sejm wniosek odrzucił. Teraz rozpatrujemy 99. poprawkę. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 99., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Przechodzimy do rozpatrzenia poprawki 100. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z państwa jest za jego przyjęciem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Kto z państwa jest za jego przyjęciem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 320. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 323. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Rozpatrujemy 324. wniosek mniejszości. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 325. wniosek mniejszości. Głosujemy.

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę przyjął. Rozpatrujemy 102. poprawkę. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 102., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Rozpatrujemy 103. poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 103. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Rozpatrujemy 104. poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 104. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął. Kto z państwa jest za jego przyjęciem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Rozpatrujemy 105. poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 105. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Głosowało 431 posłów. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Rozpatrujemy 327. wniosek mniejszości. wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Kto z państwa jest za jego przyjęciem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Rozpatrujemy 329. wniosek mniejszości. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Rozpatrujemy 106. poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 106. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Rozpatrujemy 107. poprawkę do załącznika nr 6. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki 107., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przechodzimy do rozpatrzenia 108. poprawki do załącznika nr 12. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z państwa jest za przyjęciem 108. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przed tym głosowaniem chciałabym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim parlamentarzystom, paniom i panom posłom, za prace nad ustawą budżetową, za wielogodzinne dyskusje, za bardzo merytoryczną, dobrą, rzetelną dyskusję w Komisji Finansów Publicznych, ale również w innych komisjach, gdzie te prace w bardzo aktywny sposób się toczyły. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo! Ustawa budżetowa, która przedłożona została Wysokiej Izbie, a także przeszła przez ten pełny cykl prac tutaj, w Sejmie, w parlamencie, łącznie ze wszystkimi poprawkami, została przygotowana z poszanowaniem wszystkich norm legislacyjnych zarówno prawa krajowego, jak i unijnego. Jest to budżet, który zapewnia niezbędną stabilność finansów publicznych, budżet, który jest budżetem inkluzywnym i zawierającym impulsy prorozwojowe. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za prace nad ustawą budżetową. Jestem przekonana, że jest to budżet, który będzie dobrze służył Polsce. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3021, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany w innych przepisach i załącznikach do ustawy budżetowej. Zarządzam 15-minutową przerwę i zwołuję Konwent Seniorów w ciemnym saloniku.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pani Wanda Buk przedstawi uzasadnienie projektu ustawy. Bardzo proszę. Szanowne Panie i Szanowni Panowie Posłowie! Mam przyjemność zaprezentować dzisiaj projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji, który państwu dzisiaj przedkładamy, wprowadza przede wszystkim przepisy mające na celu zwiększenie efektywności gospodarowania widmem radiowym i zapewnienie wzrostu zainteresowania wdrażaniem na rynku telekomunikacyjnym najnowocześniejszych technologii. Kwestia gospodarowania zasobami, które są dobrem dość rzadkim, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju całego rynku telekomunikacyjnego. Wprowadzane zmiany wyposażają prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w narzędzia niezbędne do prowadzenia skutecznej i efektywnej działalności regulacyjnej w obszarze widma radiowego. Projekt zawiera ponadto regulacje dostosowujące przepisy krajowe do wynikających z dyrektyw regulacji unijnych.

W projekcie nie wprowadzono zmiany systemowej, nie wprowadzono reshufflingu jako takiego.

Ponadto zgodnie z proponowanym tekstem zmiany ustawy wprowadza się możliwość wydania przez ministra cyfryzacji harmonogramu rozdysponowania częstotliwości.

Stąd też propozycja wdrożenia harmonogramu, który będzie poniekąd miał za zadanie domknięcie systemu rozdysponowywania widma. W zakresie postępowania selekcyjnego szczególną uwagę należy zwrócić na regulacje mające na celu usprawnienie prowadzonych przez prezesa UKE postępowań selekcyjnych.

Mają one na celu zabezpieczenie postępowania przed niepożądanymi zachowaniami jego uczestników.

Nowelizacja ponadto wyposaża regulatora rynku w narzędzia umożliwiające elastyczne kształtowanie warunków uczestnictwa w aukcjach i przetargach tak, aby można było zapewnić taką dystrybucję zasobów częstotliwości, która będzie wspierać równoprawną konkurencję uczestników rynku telekomunikacyjnego. Nowelizacja wprowadza także możliwość ogłoszenia przez prezesa UKE procedury selekcyjnej na zasoby częstotliwości, które są w danej chwili zajęte, ale w stosunku do których prezes UKE posiada informacje, kiedy będą dostępne w przyszłości. To rozwiązanie zapewni prezesowi UKE efektywne i ciągłe wykorzystywanie częstotliwości.

Stąd prawidłowym podejściem powinno być jak najbardziej efektywne wykorzystywanie tych częstotliwości i niedoprowadzenie do tego, aby widmo nie było użytkowane.

Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Do zabrania głosu w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość poproszę pana posła Krzysztofa Kubowa. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3116. Prawo telekomunikacyjne dotyczy przepisów z zakresu gospodarowania częstotliwościami, urządzeń radiowych i opłat za częstotliwości. Nowe przepisy dostosowują także polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Zmiany są związane z koniecznością zwiększenia efektywności gospodarowania widmem radiowym, a w szczególności zmierzają do zapewnienia wzrostu zainteresowania wdrażaniem na rynku telekomunikacyjnym nowych technologii. W projekcie ustawy zaproponowano m.in.: rozszerzenie katalogu przypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym. Jedną z ważniejszych zmian, które zaproponowano, są przepisy dające możliwość zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz czy też usprawnienie postępowania związanego z rezerwacją częstotliwości. Nowelizacja umożliwia ministrowi cyfryzacji określenie takiego harmonogramu rozdysponowania niektórych zasobów częstotliwości, aby można było realizować politykę państwa związaną z gospodarką częstotliwościami. Jednocześnie w nowelizacji ustawy zaproponowano modyfikację zasad przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, w tym w szczególności wprowadzenie dodatkowego warunku odmowy dokonania przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej takiego przedłużenia oraz umożliwienie prezesowi UKE ogłoszenia z własnej inicjatywy przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości nie tylko w przypadku posiadania wiedzy o zainteresowaniu zasobami częstotliwości, które są już dostępne. Umożliwiono także prezesowi UKE, w drodze decyzji, zmianę przydzielonych rezerwacji częstotliwości w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Proponowane rozwiązania mają służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Do realizacji tego niezbędne są zmiany w przepisach prawa, dlatego w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość proszę Wysoką Izbę o przyjęcie omawianego projektu ustawy.

Pani Minister! Wysoka Izbo! Dzisiaj trzeba powiedzieć wprost, że również telekomunikacja jest jednym z krwiobiegów gospodarki, dlatego dobre przygotowanie prawa w tym zakresie jest niezwykle istotne. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka najważniejszych kwestii, które zostały w tej ustawie zawarte.

Jeśli chodzi o narzędzia, które zostały przekazane tym projektem m.in. prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, to jest to umożliwienie cofnięcia lub zmiany rezerwacji częstotliwości w związku z wykonywaniem aktów prawnych Unii Europejskiej.

To ma właśnie temu służyć, aby unikać takich sytuacji. Jeśli chodzi o kwestie, które wzbudzają wątpliwości w tej ustawie, to jest ich kilka.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej byłby wówczas związany wytycznymi Ministerstwa Cyfryzacji, a to może naruszać przede wszystkim jego niezależność i zapisy dyrektywy europejskiej w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej. W tej dyrektywie państwa członkowskie zostały zobowiązane do zapewnienia niezależności krajowych organów regulacyjnych, zgodnie z zasadą rozdziału funkcji regulacyjnej i funkcji operacyjnej.

Tak więc kierunek generalnie jest słuszny, natomiast pewne kwestie należy wyjaśnić.

Pojawiają się informacje, że minister skłania się [[Dzwonek]] ku temu, aby było to konsorcjum, w którym będzie podmiot państwowy wraz z operatorami.

Bardzo proszę. Pani Minister! Jeżeli chodzi o zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne oraz w niektórych innych ustawach, informuję, że oczywiście mamy pewne obiekcje, jeżeli chodzi o niezależność Urzędu Komunikacji Elektronicznej od Ministerstwa Cyfryzacji, ale będziemy przyglądać się pracom, zwłaszcza na etapie drugiego czytania. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana posła Kazimierza Kotowskiego, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów, do przedstawienia stanowiska w imieniu klubu. Pani Minister! Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów jest za kontynuacją prac nad przedstawionym rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne, zawartym w druku nr 3116. Jest to naszym zdaniem pójście w kierunku, który jest oczekiwany.

Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, niemniej jednak poza tą częścią, gdzie znajdują się te odniesienia i uzupełnienia, te zapisy dotyczące aktualizacji, znajdujemy szereg zmian, szereg zapisów, które wychodzą poza tę regulację.

Uważamy, że jest to dobre, normalne, że potencjał, który mieści się w tym obszarze, powinien być wykorzystany właściwie. Powinniśmy patrzeć do przodu, powinniśmy przewidywać - i umieć wyjść im naprzeciw - te zdarzenia czy konsekwencje wydarzeń gospodarczych, aby w tym obszarze nie uczyć się od tych, co będą przed nami, a wykorzystać potencjał, który mamy, tak jak w przypadku Internetu kolejnej generacji. Jesteśmy za kontynuacją prac. Dziękuję panu posłowi. W imieniu klubu Nowoczesna głos zabierze pan poseł Mirosław Suchoń. Bardzo proszę. Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Nowoczesna w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, ujętego w druku nr 3116. Szanowni Państwo! Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu, generalnie rzecz ujmując, realizację prawa europejskiego, poprawne wdrożenie dyrektyw.

Oczywiście przedstawiony projekt ustawy niejako wychodzi naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej. Otrzymaliśmy bardzo pozytywne ogólne stanowiska dotyczące kierunku przewidzianego w projekcie ustawy. Po analizie muszę przyznać, że zgadzamy się z tym, że przepisy, które zostały zaproponowane, zmierzają we właściwym kierunku. Oczywiście jest to związane z rozwojem sieci inteligentnych, z rozwojem sieci 5G czy uruchomieniem tego nowego rozwiązania. Jak najbardziej popieramy takie działania, które prowadzą do stworzenia warunków umożliwiających lepszą gospodarkę częstotliwościami, i wytyczenie takich kierunków, które odpowiadają współczesnym wymaganiom.

Nasze wątpliwości wzbudził również przepis, który zakłada usunięcie regulacji przewidujących opłatę za wzrost wartości częstotliwości w przypadku zmiany rezerwacji. Tutaj rzeczywiście możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której niejako przypadkowo ktoś, kto bierze udział w tej, powiedziałbym, walce rynkowej o częstotliwości, stanie się beneficjentem ponad to, co zostało zadeklarowane.

W związku z przedstawionymi przeze mnie wątpliwościami wnoszę o skierowanie projektu do dalszych prac w komisji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań posłanek i panów posłów chce się.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Przepisy związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości wymagają nowelizacji ze względu na występujące nieprawidłowości.

W związku z powyższym Koło Poselskie Wolni i Solidarni jest za rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Dziękuję. W tej części głos zabierze jeszcze poseł Robert Majka, poseł niezrzeszony. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie!

Mianowicie: Czy pan premier w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej zlecił badania i przygotowanie ekspertyzy naukowej na temat wprowadzenia na terenie państwa polskiego technologii 5G? Następne pytanie: Czy premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej pan Mateusz Morawiecki zapoznał się oraz poinformował prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr. prawa Dudę o planowanym wdrożeniu w Polsce w życie technologii 5G oraz o jej wpływie na życie i zdrowie Polek i Polaków, mając na uwadze przytoczony przeze mnie cytat ze stanowiska Rady Europy z 2011 r. z rezolucji 1815?

Cztery: Czy premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej pan Mateusz Morawiecki bierze na siebie osobiście odpowiedzialność za możliwość stosowania technologii 5G w celu realizacji obowiązującej ustawy 1066 na terenie państwa polskiego przeciw narodowi polskiemu?

Dziękuję panu posłowi. Zapraszam pana posła Arkadiusza Marchewkę, klub Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, do zadania pierwszego pytania. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo!

Więc chciałbym zapytać panią minister, na jakim etapie są negocjacje z Rosją dotyczące uwolnienia tego pasma, bo bez tego oczywiście Internet piątej generacji nie będzie mógł funkcjonować. To pierwsze pytanie. Jaki jest rozważany kierunek w związku z przeprowadzeniem aukcji czy też przetargów na te częstotliwości? Czy jest taka możliwość, że w ogóle tych przetargów nie będzie, co sprawi, że również do kasy państwa [[Dzwonek]] nie wpłyną środki finansowe w tym zakresie? W jaki sposób to będzie przeprowadzane i kiedy - czy 2020 r. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Chciałbym spytać o skutki finansowe tej ustawy. W ustawie zapisane są kwoty dla budżetu państwa, które budżet państwa będzie mógł wydać w ciągu najbliższych 10 lat. Są to środki podzielone właściwie równo na ministra cyfryzacji i na urząd komunikacji elektronicznej i to specjalnie nie budzi wielkich emocji. Nie ma środków po stronie dochodów. Tu jest sytuacja odwrotna. Jednostki samorządu terytorialnego mają wydatki, ale nie mają dochodów. Mają wydatki z tytułu wydawania opłaty skarbowej, natomiast z tego tytułu nie należą im się żadne środki. Czy pani minister nie uważa, że jednak samorządy terytorialne poniosą jakieś koszty, które powinny być im zrekompensowane? Zapraszam pana posła Sylwestra Chruszcza, Wolni i Solidarni. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Właściwie miałem takie samo pytanie jak mój przedmówca.

Dziękuję. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Minister! Niestety nie skonsultowałem swojego pytania z moimi poprzednikami, bo jest nieco podobne. Jeśli tak, to na jaki okres i czy zostały wprowadzone mechanizmy zabezpieczające te środki? Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Chcę zapytać, czy rząd jest pewien, że umożliwienie odgórnego, z urzędu zmieniania koncesji radiowo-telewizyjnych na rzecz dobrych kilkuset nadawców radiowych i kilkudziesięciu nadawców telewizyjnych w Polsce, spowodowane chęcią zajęcia ich częstotliwości przez technologię 5G, nie spowoduje ograniczenia dostępu do wolności słowa w Polsce, a więc czy rzeczywiście jest tak, że zapewnienia o tym, że równorzędne częstotliwości przyznawane tym podmiotom nie spowodują zakłócenia na rynku radiowo-telewizyjnym ani dostępu do informacji, a także nie naruszą praw koncesjonariuszy, którzy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji uzyskali w ciągu ostatnich 30 lat koncesję na nadawanie radiowo-telewizyjne. I zapraszam panią poseł Zofię Czernow, Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, do zadania pytania. Pani Minister! Również chciałam zapytać o finanse, ale nieco inaczej. Zgodnie z projektem ustawa wejdzie w życie w ciągu 30 dni od daty jej ogłoszenia, tymczasem w projekcie budżetu na cały ten rok, czyli na trzy kwartały, nie ma żadnych środków finansowych na realizację tej ustawy. Aby ustawę można było realizować, konieczne jest zatrudnienie wysokiej klasy ekspertów, a także wyposażenie ich w odpowiednie urządzenia najnowszej generacji.

Jestem po prostu zaskoczona, że nie zabezpieczamy realizacji ustawy. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Pani Minister! Po pierwsze, z czego konkretnie wynika dystans 500 m, jeżeli chodzi o odległość od urządzeń pomiarowych?

I po drugie, kiedy tak naprawdę.

Przecież nie mamy jeszcze żadnych uzgodnień z sąsiadami, które pozwoliłyby na to, żeby zacząć ją realizować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Premier ostatnio powiedział, że jest zwolennikiem budowy jednej sieci. Czy Ministerstwo Cyfryzacji ma plan, koncepcję, strategię, jaką sieć 5G chce budować, czy nie?

Pan poseł Marek Wójcik, Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Chciałbym zapytać o przewidzianą w ustawie strefę ochronną wokół urządzeń pomiarowych UKE. Zgodnie z projektem operatorzy telekomunikacyjni nie będą mogli instalować nadajników w promieniu 500 m od urządzeń pomiarowych.

Ich obecnie nie jest dużo.

Natomiast jeżeli wprowadzimy zakaz instalowania nadajników 5G właśnie w tym miejscu, to spore osiedla w Siemianowicach, również w Katowicach będą właściwie pozbawione możliwości korzystania z tych usług. Dlatego bardzo proszę o podanie informacji, z czego wynika ten zakaz i czy państwo przeprowadzaliście jakieś nowe analizy dotyczące konieczności wprowadzenia tej strefy ochronnej. Bardzo proszę. Pani Minister! Wysoka Izbo! Pani minister, chciałem zapytać o kwestię centrów dużych miast.

Druga kwestia dotyczy art. 118 ust. 2c, który wprowadza bardzo rygorystyczny przepis w zakresie odpowiedzialności karnej za błąd w informacji zawartej w ofercie składanej w ramach aukcji lub przetargu.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Rozmawiamy o pięknych, ambitnych planach budowy sieci 5G. W tym kontekście pojawiają się pytania o możliwość wystąpienia białych plam. A co z tymi białymi plamami, które dzisiaj mamy, które dzisiaj utrudniają i uniemożliwiają obywatelom korzystanie z telefonów komórkowych?

Czy ministerstwo chce stawiać własne maszty, czy chce budować jedną, jednolitą sieć, czy chce, być może, stworzyć jakiś system zachęt dla operatorów komórkowych albo operatorów tych masztów, żeby Polska faktycznie była państwem w 100% [[Dzwonek]] pokrytym zasięgiem sieci komórkowej, nawet 3G, żeby ona po prostu była? Wysoka Izbo! Należy kontynuować prace nad tym projektem, aby to prawo było zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, niemniej jednak należy doprecyzować niektóre zapisy w taki sposób, abyśmy mogli dobrze wykorzystać potencjał Internetu.

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Minister!

Bardzo proszę.

Nie jest to ustawa, która wprowadza technologię 5G.

Obawy społeczne, o których wspominał pan poseł, jak rozumiem, dotyczą tego obszaru fizyki.

Sieć 5G to jest tak naprawdę kolejny etap rozwoju sieci telekomunikacyjnej, tu nie będzie nic budowane od zera, operatorzy telekomunikacyjni naturalnie będą wykorzystywać tę infrastrukturę, którą już dzisiaj posiadają.

Siedemsetka jeszcze nie jest ostatecznie przeznaczona, ale faktycznie zaraz będzie.

To jest technologia.

Natomiast w kolejnych latach w ustawie budżetowej już zostaną przewidziane środki na dodatkowe etaty.

Należy też podkreślić, że w miastach - bo mówimy tutaj przede wszystkim o miastach - ta sieć jest tak gęsta, że można ją wykorzystywać alternatywnie. Dokładnie na odwrót, niż zostało tutaj wskazane - można wykorzystywać komórki o małej mocy, które tym bardziej nie będą zakłócać urządzeń UKE. Dziękuję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 3116, do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3045) Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pan Michał Dworczyk przedstawi uzasadnienie projektu.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw. Projekt jest istotny ze względu na podjętą w nim próbę uporządkowania ważnej dla opinii publicznej kwestii odpowiedniego uhonorowania osób, które ze względu na swoją działalność, wybitne osiągnięcia i ponadprzeciętną postawę społeczną zasługują na otrzymanie specjalnej nagrody o charakterze finansowym. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają wskazanym ministrom na przyznawanie nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia, niemniej jest to mechanizm dalece niewystarczający. Po pierwsze, należy wskazać, że przepisy dotyczące przyznawania nagród specjalnych powstawały na przestrzeni wielu lat i w konsekwencji charakteryzują się nie tylko niespójnością przesłanek ich przyznawania, ale także znaczną rozpiętością kwot, jakie na te nagrody mogą być przeznaczane.

Po drugie, w myśl obecnych przepisów niezwykle trudne, a czasami wręcz niemożliwe jest uhonorowanie osiągnięć o charakterze ponadstandardowym i interdyscyplinarnym, czyli niemieszczących się w żadnym sztywnym systemie działów administracji rządowej, oraz osiągnięć tak wybitnych i niepowtarzalnych, że zasługują na szczególne uhonorowanie. Przedstawiany Wysokiej Izbie projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom w zakresie należytego, godnego i adekwatnego uhonorowania osób, które mogą poszczycić się szczególnie spektakularnymi osiągnięciami. Projekt daje prezesowi Rady Ministrów możliwość przyznania w takich przypadkach nagrody specjalnej, nagrody, która będzie mogła być udzielona niezależnie od innych form uhonorowania danego osiągnięcia, nagród przydzielonych przez właściwego ministra.

Z kolei przez przewidziane w projekcie ustawy finansowanie przyznanej nagrody specjalnej z rezerwy ogólnej budżetu państwa zapewniona zostanie pełna transparentność całego procesu. Przyznanie nagrody specjalnej będzie bowiem każdorazowo wymagało wydania przez prezesa Rady Ministrów stosownego zarządzenia, łączna zaś wysokość nagród specjalnych udzielanych w danym roku limitowana będzie wysokością środków pozostałych w ramach rezerwy ogólnej, po uprzednim uwzględnieniu wszystkich innych potrzeb z niej finansowanych. Nie budzi wątpliwości to, że wybitne osiągnięcia wymagają szczególnego uhonorowania. W obecnym systemie prawnym jest to nie tylko znacznie utrudnione, ale w wielu przypadkach wręcz niemożliwe. Dzięki przedłożonej Wysokiej Izbie ustawie o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw stanie się możliwe odpowiednie uhonorowanie najwybitniejszych osiągnięć i postaw społecznych, które, z jednej strony, rozsławiają nasz kraj poza granicami, takich jak dokonania sportowców, z drugiej zaś strony, stanowią doskonały przykład do naśladowania dla wszystkich Polaków. Wysoka Izbo! Pani Marszałek! Dziękuję panu ministrowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość wystąpi pan poseł Piotr Kaleta. Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3045.

Proszę Państwa! To dobra ustawa, ustawa, która w moim najgłębszym przekonaniu mogłaby być wprowadzona już dawno, ponieważ, cokolwiek by mówić, jeżeli chodzi o osobę nagradzaną przez prezesa Rady Ministrów, przez premiera rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, to ma to niewątpliwy wymiar społeczny, ale także wymiar, który polega na tym, że jest to niewątpliwy zaszczyt dla tych osób, które są nagradzane. W związku z tym myślę, że mówienie dzisiaj o kwestiach łączących się ze sprawami finansowymi, o tym, o jakich nagrodach byśmy mieli tutaj wspominać, w jakich wysokościach, niekoniecznie jest uprawnione, ponieważ zdawać sobie musimy sprawę z tego, że mamy tutaj do czynienia z wszelakimi rodzajami postaw społecznych, kulturalnych, sportowych, które trudno jest jednoznacznie oceniać.

Niejako prosi się to o to, żeby za te chwile wzruszeń, za te chwile naszej narodowej dumy również chociażby w sposób symboliczny te osoby zostały nagrodzone. Jestem o tym głęboko przekonany, że ta ustawa znajdzie poparcie w Wysokiej Izbie - również innych klubów - ponieważ nie jest ona ustawą, która powinna budzić czy budzi kontrowersje. Tak po prostu powinno w naszym kraju być od dawna. W związku z tym proszę państwa, nie przedłużając wystąpienia, bo wydaje mi się, że ta ustawa ma charakter oczywisty i pewnie będzie debatowana również w innych miejscach, tak żeby ją jeszcze w sposób należyty dopracować, chciałbym prosić Wysoką Izbę o poparcie. Dziękuję panu posłowi. W imieniu klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska głos zabierze pan poseł Grzegorz Lipiec.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Ministrów - tak ładnie się to nazywa - jest generalnie ustawą o dodatkowych możliwościach premiera w roku 2019, czyli o przyznawaniu rozmaitych nagród specjalnych w tych obszarach, w których do tej pory robili to ministrowie.

A premierów przecież nasz kraj miał już bardzo wielu i akurat nie wiadomo, dlaczego jeszcze tego uprawnienia premier nie ma. Przecież bardzo łatwo można sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało w praktyce.

To przecież ministrowie mają cały aparat urzędniczy, mają względnie największą wiedzę o tym, kogo można uhonorować, komu te nagrody można wręczyć, mają odpowiedni aparat weryfikacyjny.

No chyba nikt nie ma wątpliwości, my również ich nie mamy. To dziesiątki, a może nawet setki dodatkowych zdjęć rozmaitych zadowolonych naukowców, sportowców czy osób aktywnych w obszarach kultury, którym dobry premier będzie wręczać taką czy inną nagrodę, bo przecież to on jest twarzą czy był twarzą, będzie twarzą kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Czy naprawdę ktoś na tej sali myśli, że nie może być osobą, która w obszarze sportu przyznaje nagrody, np. minister sportu, np. pan minister Bańka, czy też w obszarze kultury i nauki, gdzie dwóch wicepremierów się tym zajmuje. A więc premier w roku wyborczym będzie mógł wszystko, przecież może dogadywać się z premierem Glińskim i Gowinem. W związku z tym trudno mi sobie wyobrazić, że akurat oni mu się jakoś szczególnie sprzeciwią. I nie wiem, czemu akurat mamy obciążać go tą dodatkową pracą, a wiemy przecież, że premier jest osobą bardzo zapracowaną i ma dużo swoich obowiązków. Może chodzi o pokazanie, kto tu rządzi, żeby jeszcze ministrom coś odebrać i jeszcze robić coś po swojemu. Ona jest bardzo krótka.

Na pewno klub Platformy Obywatelskiej na posiedzeniu komisji będzie wspierał rozwiązania, które będą ułatwiać przecież życie tym najwybitniejszym spośród Polaków. Ale nie widzimy jakiegoś szczególnego powodu, żeby akurat w roku 2019 trzeba było obarczać premiera jakimiś szczególnymi, nowymi obowiązkami, bo przecież ma co robić, jest dużo pracy w naszym kraju i nie ma takiego szczególnego powodu, żeby tego nie mógł robić odpowiedni minister, a przecież trudno uwierzyć, że minister nie będzie realizować tego, co uzgodni ze swoim prezesem Rady Ministrów.

I drodzy państwo, mówimy o ustawie, która ma przyznać uprawnienie prezesowi Rady Ministrów do przyznawania specjalnej nagrody. I znów państwo w sprytny sposób operujecie słowem, bo z jednej strony mówicie o wybitnych zasługach, o wybitnych osobistościach, ludziach sportu, ludziach kultury, wynalazcach, naukowcach, o kimkolwiek, kto w szczytny sposób przyczynił się do wzmacniania naszej ojczyzny, do potęgowania jej dobrego imienia. I patrząc się w tym kierunku, wydawać by się mogło, że to jest słuszne rozwiązanie, tylko że dzisiaj ministrowie mają już uprawnienie do tego, żeby takie nagrody przyznawać. Pan poseł Kaleta mówi, że chodzi o rangę, żeby to premier przyznawał taką nagrodę. Też jest to jakiś argument. Natomiast, drodzy państwo, niestety sprawa wygląda trochę tak, że oto pan premier chce się uniezależnić od ministra, a być może chce po prostu pozbyć się ministra u swojego boku po to, żeby mógł sam tę nagrodę przyznawać, a nie być niejako obok tego, który tę nagrodę wręcza. Budzi to duże wątpliwości, ale przede wszystkim nasze wątpliwości budzi brak ograniczenia, brak określenia, jaka ma być wysokość tych nagród. Pan minister Dworczyk mówił o tym, że suma nagród nie może przekroczyć tej części budżetowej określonej jako rezerwa ogólna pomniejszona oczywiście o te wszystkie elementy składowe wyszczególnione w rezerwie ogólnej, przeznaczone na realizację różnych projektów, inwestycji itd. Ale, panie ministrze, to wciąż są kolosalne pieniądze. Ja oczywiście, być może w swojej naiwności, ale jednak wierzę w to, że pan premier, dbając de facto o swój wizerunek, nie roztrwoni kilku miliardów złotych, przeznaczając je na nagrody, bo to byłoby po porostu nieprzyzwoite. Ale czy nie warto wypracować pewnych rozwiązań granicznych, takich, które jednak nakładałyby pewne ograniczenia? Drodzy państwo, jak dobrze wiemy, i nie jest to absolutnie zarzut, pan premier jest człowiekiem zamożnym, to dobrze, ale nie może być tak, że oto Mateusz Morawiecki czy każdy inny, przyszły, następujący po nim premier będzie mógł swobodnie dysponować pieniędzmi tak naprawdę płaconymi przez obywateli, należącymi do obywateli, ponieważ ani premier Morawiecki, ani żaden wcześniejszy premier i późniejszy, następujący po nim, nie ma żadnych swoich pieniędzy. Rząd nie ma swoich pieniędzy, jeżeli mówimy o pieniądzach budżetowych. Budżet tworzy się z podatków, tworzy się z ciężkiej pracy obywateli. Dlatego bardzo bym chciał, aby te pieniądze, które Polacy z trudem wypracowują, a które państwo z łatwością odbierają w formie podatków, nie były z równą łatwością rozdysponowywane, jak się komu żywnie podoba. Żeby jednak nie było, że są to same złe rozwiązania, zwróciliśmy uwagę, ja zwracam uwagę, na jedno bardzo dobre rozwiązanie, które może być pewnego rodzaju światełkiem, taką jaskółką. Mianowicie jest w tym krótkim projekcie ustawy taki zapis, że ta nagroda będzie zwolniona z podatku dochodowego. To słuszne rozwiązanie oczywiście, podobnie zresztą jak czymś słusznym jest niepobieranie po raz drugi podatku od emerytury, ale to inny projekt. Natomiast, drodzy państwo, zwróćcie uwagę: być może to jest właśnie kierunek, w którym warto iść, tak żeby likwidować te wypłaty, które są objęte podatkiem dochodowym, i rozszerzyć zakres tych wypłat, które nie są objęte podatkiem dochodowym, bo tak naprawdę im więcej pieniędzy pozostanie w kieszeni obywateli, tym większy będzie cash flow, czyli obrót pieniądza w gospodarce, a gospodarka rozwija się głównie poprzez właśnie obrót pieniądza, zakupywanie usług i ich świadczenie. Natomiast, drodzy państwo, kończąc - niewątpliwie projekt wymaga dopracowania, dlatego będziemy rekomendować, żeby po prostu został [[Dzwonek]] skierowany do komisji, gdzie pewne ramy, ograniczenia zostaną wypracowane, zastosowane, bo chodzi o pieniądze obywateli. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów głos zabierze pan poseł Łopata. Ale zanim to się stanie, pozwoli pan, panie pośle, że przywitam członków Stowarzyszenia Aktywni Razem z miejscowości Ludomy, którzy przyjechali [[Oklaski]] na zaproszenie pana posła Krzysztofa Paszyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszystkiego dobrego. Witamy serdecznie. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów pragnę zaprezentować nasze stanowisko, naszą opinię co do projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw. Wysoka Izbo!

Zmiany zmierzają do umożliwienia właśnie prezesowi Rady Ministrów, premierowi przyznawania osobom fizycznym w szczególnie uzasadnionych przypadkach - te przypadki zostały tu wymienione, to są wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe czy też z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - nagród specjalnych.

Jesteśmy dzisiaj już trochę dalej.

Wysoki Sejmie! Tak jak zaznaczyłem na wstępie, potwierdzam też teraz w imieniu klubu PSL - Unii Europejskich Demokratów: jesteśmy za przyjęciem uregulowań zawartych w tym projekcie ustawy. Dziękuję. I zapraszam na mównicę panią poseł Paulinę Hennig-Kloskę, klub Nowoczesna, celem przedstawienia stanowiska w imieniu tego klubu. Panie i Panowie Posłowie!

Bo to, że pan premier chciałby dołączyć do grona ministrów, którzy takie nagrody mogą przyznawać, wydaje się rzeczą zasadną.

Ale biorąc pod uwagę, tak jak powiedziałam, tryb procedowania nad ustawą, a także datę jej wejścia w życie, zaraz zastanawiam się, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, czy pan premier przyznał już jakieś nagrody, do których przyznania uprawnień nie posiadał, albo komu pan prezes już obiecał, nie wiedząc, że nie ma takiej kompetencji. Pamiętamy powrót siatkarzy z ostatnich mistrzostw i wiemy, że takie obietnice z ust pana premiera padły.

Tak jak pan premier wcześniej jeździł po regionach, obiecując inwestycje, pod warunkiem że Prawo i Sprawiedliwość w danym województwie czy w danej miejscowości wygra wybory, tak, mam wrażenie, dzisiaj mamy do czynienia z bardzo podobną potrzebą, tylko szukacie sposobu, chodzi o to, jakie narzędzia dać panu premierowi, żeby jako twarz kampanii Prawa i Sprawiedliwości mógł jeździć po województwach, po miastach, po wsiach i przyznawać nagrody. Pan mówi, że mamy tu ograniczenie rezerwy ogólnej, ale dobrze wiemy - akurat jestem posłem pracującym w Komisji Finansów Publicznych - że ta rezerwa ogólna jest wyjątkowo duża w tym roku. Takie obawy już zgłaszaliśmy w trakcie prac w Komisji Finansów Publicznych, że z tej rezerwy ogólnej będą brane pieniądze po to, żeby obiecać kolejne inwestycje, korumpując w ten sposób obywateli albo ucząc ich takiego myślenia, że oto w zamian za poparcie w danym regionie rząd wybuduje to właśnie tu szkołę, to właśnie tu szpital, to właśnie tu nową halę. Nie, tak się nie da rządzić państwem, bo w gruncie rzeczy wszyscy obywatele na ten budżet się składają, niezależnie od regionu, miasta czy wsi, w których mieszkają. Rząd nie ma prawa rozdawać pieniędzy publicznych - do których się nie dokłada, na które składają się obywatele - według jakiegoś własnego, nikomu nieznanego albo dobrze znanego harmonogramu i zasad. Powinien je dzielić równo między wszystkich Polaków, bo wszyscy Polacy równo, tak jak powiedziałam, na budżet się składają. Tak że oczywiście jesteśmy za tym, żeby nad tą ustawą dalej pracować w komisji właściwej, natomiast, tak jak powiedziałam, te wątpliwości są. Zasada, że prawo nie działa wstecz, dzisiaj już was nie obowiązuje, mało tego - to, że prawa nie tworzy się wstecz, również, jak widać po tej ustawie, was nie obowiązuje. I to już jest dla nas rzecz nie do zaakceptowania. Zapraszam panią poseł Małgorzatę Zwiercan, koło Wolni i Solidarni, w celu przedstawienia stanowiska w imieniu tego właśnie koła. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw. Nie mam wątpliwości, że Polacy są narodem niezwykle utalentowanym, i to na wielu polach; że dzięki konsekwencji, determinacji i ciężkiej pracy potrafimy wznosić się na wyżyny i osiągać stawiane sobie cele, często niezwykle trudne. Dlatego fakt, że nasi reprezentanci doceniani są w wielu dziedzinach na arenie międzynarodowej, zdobywają złote medale na olimpiadach czy mistrzostwach świata, w ogóle mnie nie dziwi, a przepełnia mnie narodową dumą. Ważne jest jednak, by te osiągnięcia, oprócz uznania i wdzięczności rodaków, w sposób adekwatny wynagradzane były materialnie. W moim przekonaniu polskie państwo powinno pokazać, że docenia dokonania i sukcesy swoich przedstawicieli. Wedle regulacji zawartych w omawianym projekcie premier będzie mógł, za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe czy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii odpowiedniego ministra, przyznawać nagrody specjalne. Panie Ministrze!

Wszyscy wiemy, że to był bardzo duży triumf, niemniej prawo nie działa wstecz. Wysoka Izbo! Projekt ten jest potrzebny i nie powinien budzić niczyjego sprzeciwu. Ufam, że taka nagroda za ponadprzeciętne rezultaty jeszcze bardziej będzie motywować Polaków do skuteczniejszego własnego rozwoju, jeszcze bardziej wytężonej pracy i zdobywania kolejnych szczytów. Koło Wolni i Solidarni popiera zaproponowane rozwiązania. Dziękuję. Czy ktoś z pań posłanek i panów posłów chce jeszcze wpisać się na listę osób, które zamierzają zadać pytanie w tym punkcie? Zamykam więc listę. Zapraszam pana posła Marka Wójcika, klub Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, do zadania pierwszego pytania. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Słuchałem uważnie pana ministra i mam wrażenie, że pan minister przedstawiał argumentację dotyczącą chyba innej ustawy niż ta, nad którą tutaj procedujemy, dlatego że pan minister mówił o porządkowaniu przepisów, tymczasem w tej ustawie nie ma słowa o porządkowaniu przepisów, bo państwo po prostu, jeśli chodzi o istniejące przepisy i możliwość przyznawania nagród przez ministrów, dokładacie kolejną nagrodę - nagrodę premiera.

Chciałbym również zapytać, czy przewidujecie państwo jakąś maksymalną wysokość nagrody i czy fakt przyznania nagrody przez prezesa Rady Ministrów będzie wykluczał możliwość przyznania nagrody specjalnej tej samej osobie za to samo osiągnięcie przez ministra, dlatego że dziś to minister przyznaje nagrodę, natomiast państwo proponujecie, żeby w przypadku nagrody specjalnej [[Dzwonek]] jeszcze pytać o opinię tego ministra resortowego, który przecież też ma własne uprawnienie do przyznawania tej nagrody.

Bardzo proszę. Dziękuję. Mam pytanie właśnie o te ramy: Jakie będą zasady przyznawania tych nagród? To po pierwsze. Pytam, żeby to było jasne, transparentne, jawne. To jest pierwsza, podstawowa sprawa. Kolejna kwestia dotyczy tego, czy będzie również jakieś ograniczenie o charakterze ogólnym, bo ograniczenie do poziomu rezerwy ogólnej w budżecie państwa - sami państwo przyznacie - jest chyba trochę zbyt dużą frywolnością i swobodą w podejściu do wydatkowania jednak publicznych pieniędzy. Absolutnie nie jesteśmy przeciwni temu, żeby nagradzać wybitne postacie czy kultury, czy sportu, czy nauki, natomiast bardzo byśmy chcieli, żeby zostały ustalone takie ramy prawne, które będą, że tak powiem, zachowywały racjonalność w wydatkowaniu [[Dzwonek]] środków publicznych, czyli pieniędzy należących do obywateli. Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Bardzo dobrze się stało, że ta regulacja jest. I to nie jest nagroda wicewójta, wicestarosty, wiceburmistrza czy wiceprezydenta. Są to nagrody prezydenta, wójta, starosty. Natomiast chciałem się zapytać o coś takiego, bo usłyszałem: naukowcy, sportowcy, z zakresu kultury, dziedzictwa. Mówimy tu o olimpijczykach, sportowcach. Chodzi mi o TOPR-owców i GOPR-owców, czyli za wybitne osiągnięcia w ratowania życia, naukowe, sportowe. Być może to jest zbyt szerokie, ale czy nie należałoby ich tu ująć? Pan poseł Piotr Pyzik,

Wysoka Izbo! Prezes Rady Ministrów będzie mógł przyznawać nagrody specjalne, a środki na te nagrody specjalne będą pochodzić oczywiście z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Jaką planuje się na ten cel sumę środków finansowych na rok 2019? Bo w uzasadnieniu ustawy czytam, że proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Tak się zagalopowaliście, żeby zdążyć w roku wyborczym, że nawet wam się daty pomyliły. Mam pytania. Kto będzie wskazywał osoby, które będą nagradzane? Jakie będą kryteria? W mojej ocenie każdy minister ma takie kompetencje nagradzania wybitnych osób, więc zbyteczne jest obciążanie prezesa Rady Ministrów dodatkową pracą, bo przecież jest tak bardzo [[Dzwonek]] zapracowany. Panie Ministrze! Wszyscy pamiętamy, że w ostatnich miesiącach Sejm przyjął ustawę, w przypadku której dokonał zwiększenia zakresu uprawnień prezesa Rady Ministrów, które może nie do końca były uregulowane. Bardzo żałuję, że wówczas nie zajęto się sprawą tych nagród, bo wtedy istniała możliwość, żeby w budżecie państwa zabezpieczyć środki na ten cel. Nie jest ona wysoka, a na pewno nie można dysponować nią od stycznia. Ona po prostu służy wtedy, kiedy ze względu na sytuacje budżetową konieczne jest sięgnięcie do tej rezerwy. Tutaj powstają wątpliwości, kto będzie zajmował się przyznawaniem nagród i jaką rangę będą miały dotychczasowe nagrody ministrów. Przecież one stracą swoją rangę. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Oczywiście trudno uciec od takiej opinii i takiego wrażenia, że jednak ten projekt ustawy, który przewiduje dodatkowe uprawnienia dla premiera, dla prezesa Rady Ministrów w postaci możliwości przyznania nagrody za osiągnięcia, które są wymienione w ustawie, jest projektem, który wpisuje się w szerszą koncepcję tworzenia takiego urzędu superpremiera, bo przecież mieliśmy już takie projekty, które pozbawiały ministrów części odpowiedzialności i przenosiły ją właśnie na premiera, w Sejmie leży projekt, który tworzy nowy fundusz, który również będzie w zasadzie w dyspozycji premiera, premier będzie mógł jednoosobowo decydować. To jest kolejny taki projekt. Muszę powiedzieć, że państwo polskie powinno doceniać wszystkie osoby, które w sposób szczególny wpisują się w te cele z uzasadnienia ustawy, natomiast państwo polskie [[Dzwonek]] to robi.

Dziękuję bardzo. Zapraszam pana posła Jarosława Gonciarza z Prawa i Sprawiedliwości do zadania kolejnego pytania. Panie Ministrze! Uważam, że kultura, przyzwoitość, szacunek przemawiają za zapisem, że prezes Rady Ministrów może przyznać nagrodę specjalną osobie fizycznej - po zasięgnięciu opinii właściwego ministra. Moim zdaniem taka opinia w tym przypadku jest zbędna. Moje pytanie: Czy konieczny jest zapis o opinii? Dziękuję. Proszę bardzo.

Wysoka Izbo!

Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Najpierw pytanie do pana ministra: Kto będzie mógł wnioskować o te nagrody?

Pani poseł z Nowoczesnej, która była łaskawa przedstawić stanowisko klubu, powiedziała coś takiego, co nie bardzo zrozumiałem.

Kolejna sprawa, dotycząca wypowiedzi posłów Kukiza. To są pieniądze rządu czy to są pieniądze Polaków?

Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Przypominam, że na tej sali powinno się raczej merytorycznie zadawać pytania, a nie obrażać posłów. także mnie, bo ja z tego klubu jestem. Bardzo proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pana Michała Dworczyka. Bardzo proszę, panie ministrze. Wysoka Izbo! Postaram się odpowiedzieć na pytania, które padły na tej sali.

Chciałoby się powiedzieć: nie wszystkich swoją miarą. Wystarczyło przeczytać uzasadnienie i metryczkę, zobaczyć, jak ta ustawa była procedowana, żeby wiedzieć, że Rada Ministrów w listopadzie ten projekt przyjęła.

Tam jest informacja, a w dodatkowych materiałach na pewno można znaleźć taką informację, że dzisiaj tylko czterech ministrów na 19 ministerstw posiada takie kompetencje, żeby przyznać nagrodę.

Dzięki projektowanej ustawie tę lukę właśnie likwidujemy.

On wziął się właśnie stąd, że projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów jesienią. To jest oczywiście słuszna uwaga.

Po raz kolejny pojawiło się takie pytanie, czy na pewno jest potrzebne to, żeby prezes Rady Ministrów mógł przyznawać takie nagrody.

To jest pewna filozofia patrzenia na rolę prezesa Rady Ministrów i w ogóle na funkcjonowanie rządu.

I wydaje mi się, że jeśli chodzi o funkcjonowanie władzy, w tym wypadku władzy wykonawczej, rządu, w tym wypadku prezesa Rady Ministrów, to też jest potrzebne minimum zaufania. Bo znowu padło w jednej wypowiedzi pytanie: Czy to będzie jawne? Każda taka nagroda jest przyznana zarządzeniem prezesa Rady Ministrów, a każde zarządzenie jest publikowane w BIP.

Proszę państwa, w rezerwie ogólnej - wystarczy spojrzeć do ustawy budżetowej - jest w tym roku chyba 250 mln zł.

I trzeba pamiętać, że ta rezerwa jest przeznaczona przede wszystkim na inne sytuacje.

O terminie wejścia mówiłem, o rezerwie ogólnej mówiłem.

Myślę, że będzie to związane ze zmianą w regulaminie funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale będzie tu chodziło o Biuro Prezesa Rady Ministrów, czyli o jedną z komórek, która opracowuje dla pana premiera materiały na co dzień.

Ostateczna decyzja i tak będzie zależała od pana premiera.

Oczywiście tak.

Na pytanie pana posła Suchonia o to, ile pieniędzy i którzy ministrowie przyznali w roku 2018 w ramach nagród resortowych, odpowiem na piśmie, bo muszę to zweryfikować. Wnioskować może każdy, natomiast decyzję ostatecznie podejmuje prezes Rady Ministrów.

Dzisiaj to Prawo i Sprawiedliwość ma większość parlamentarną, za rok, może za kilka lat, to będzie jakaś inna partia i będzie inny premier, a to narzędzie pozostanie.

Bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 3045, do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3072 i 3126) Pan poseł Jerzy Polaczek przedstawi sprawozdanie komisji. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić syntetyczne sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, który jest zawarty w drukach nr 3072 i 3126.

Wdrożenie tej dyrektywy wiąże się z potrzebą dodania nowych celów, dla których wydawane są wizy, tj. odbycia stażu oraz udziału w programie wolontariatu europejskiego, a także wprowadzenia zmian w zakresie przepisów regulujących udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, w celu prowadzenia badań naukowych, dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskie lub cudzoziemców oraz zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności. Projektowane zmiany mają również na celu uporządkowanie regulacji dotyczących korzystania przez cudzoziemców z różnych rodzajów mobilności na terenie naszego kraju, do czego nie zawsze konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy. Warto zauważyć, iż na szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nakładane są nowe obowiązki informacyjne względem komendanta głównego Straży Granicznej oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także innych państw członkowskich związane z korzystaniem z różnych rodzajów mobilności na terytorium Polski.

Wysoka Izbo!

To zjawisko polega na składaniu wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez obywateli państw trzecich, najczęściej są to państwa nieeuropejskie, np. Irak, Pakistan, Bangladesz czy Indie. Ci obywatele na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywają bardzo krótko, zazwyczaj w oparciu o wizę Schengen wydaną przez inne państwo obszaru Schengen. W związku z tym proponujemy w tej regulacji dodanie dwóch nowych przesłanek odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia odpowiednio zezwolenia na pobyt czasowy oraz pracę oraz zezwolenia w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, które będą zależne od tego, na jakiej podstawie cudzoziemiec przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w chwili złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy danego rodzaju. Chciałbym naprawdę bardzo skrótowo zasygnalizować kilka poprawek merytorycznych, które zostały przyjęte przez podkomisję nadzwyczajną, która została powołana na posiedzeniu w dniu 10 stycznia.

Ta poprawka polega na doprecyzowaniu, że z obowiązku zatwierdzania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów zostaną zwolnione uczelnie prowadzone przez Kościoły i związki wyznaniowe, ale tylko takie, których stosunek do Rzeczypospolitej Polskiej reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa. Ma to na celu zapobieżenie zagrożeniu dla bezpieczeństwa państwa wynikającemu z możliwości tworzenia się w kraju uczelni zakładanych przez działający w Polsce Kościół lub związek wyznaniowy, za pośrednictwem których o zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia na studiach będą ubiegały się osoby o poglądach bądź zachowaniu sprzecznych z zasadami porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę na poprawkę dotyczącą art. 188 ust. 2a ustawy o cudzoziemcach. Ta przyjęta przez komisję poprawka polega na doprecyzowaniu, że cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności z uwagi na to, że jest absolwentem polskiej uczelni i poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium, powinien przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych, ale na polskiej uczelni. Dotychczasowa propozycja w tym zakresie wskazywała jedynie na konieczność przedstawienia dyplomu ukończenia studiów wyższych bez tego doprecyzowania.

Zgodnie z dodawanym brzmieniem w rejestrze tym będą przechowywane informacje o zawiadomieniach, dokumentach załączonych do zawiadomień, jak również informacje o decyzjach szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o sprzeciwie. Kolejna poprawka, która jest warta odnotowania, polega na dodaniu regulacji przejściowej w art. 14 projektu. Zgodnie z tą poprawką zaświadczenia, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o cudzoziemcach, wydawane uczestnikom studiów doktoranckich w okresie od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. będą wydawane w oparciu o przepisy w brzmieniu nadanym tą ustawą z tym tylko zastrzeżeniem, że informacje w nich zawarte powinny odzwierciedlać to, że studia doktoranckie mogą być prowadzone w określonej dyscyplinie naukowej lub artystycznej. Przepis ten został ustanowiony w celu odróżnienia doktorantów będących uczestnikami studiów doktoranckich, które mogą być jeszcze prowadzone na zasadach dotychczasowych, tj. sprzed wejścia w życie

W projekcie przewiduje się opóźnienie wejścia w życie części przepisów ustanawiających kompetencje szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców do wydawania decyzji o sprzeciwie w przypadkach zawiadomień o zamiarze korzystania przez cudzoziemców z odpowiednich rodzajów mobilności. Jest to spowodowane dostrzeżoną przez rząd koniecznością przygotowania się organów administracji publicznej do tego całkowicie nowego zadania. Do tej pory polskie przepisy w zakresie wjazdu i pobytu cudzoziemców nie przewidywały funkcjonowania podobnej instytucji.

Do projektu zostały również wprowadzone poprawki o charakterze legislacyjnym oraz redakcyjnym.

Dziękuję za uwagę. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Panie i Panowie!

I zapraszam do zabrania głosu w imieniu klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska panią poseł Annę Nemś. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

W projekcie tym redefiniuje się pojęcie mobilności, określa się m.in. katalog przyczyn odmowy wydania wizy studenckiej nie tylko w przypadku uchybień po stronie kandydata, ale także w przypadku udokumentowanych złych praktyk jednostek akademickich, które mogą prowadzić do nielegalnego sprowadzania cudzoziemców do Polski.

Pewnie nie jest to czas ani miejsce, żeby o tym rozmawiać, bo to jest tylko implementacja, technicznie dobrze przygotowana, ale problem pozostaje i chciałabym zwrócić na te sprawy uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam, zgadza się. Pan poseł Józef Lassota, także Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Zostało jeszcze trochę czasu, a więc bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo!

Oczywiście projekt faktycznie jest niekontrowersyjny, bo w zasadzie jest projektem technicznym, regulującym różnego rodzaju sprawy związane z pobytem cudzoziemców, ale zastanawialiśmy się, czy faktycznie jest potrzeba aż tak szczegółowego opisu różnych detalicznych czynności w ustawie.

Może warto się pokusić o inne podejście do redagowania ustaw, nie na zasadzie przepisu instrukcyjnego. Dziękuję bardzo. A teraz już pan poseł Paweł Skutecki, klub Kukiz’15. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która jest tak naprawdę implementacją dyrektywy, nie budzi kontrowersji, bo nie powinna budzić kontrowersji.

Panie ministrze, wiem, że to nie jest w zakresie kompetencyjnym ministerstwa, którym pan zawiaduje, natomiast jest to bardziej temat dla rządu.

Co to będzie znaczyło dla polskiej gospodarki, mniej więcej wszyscy wiemy, na pewno ona się zachwieje, a nie wiadomo, czy to się nie skończy większymi problemami. I teraz mamy tylko jedną alternatywę, jedną prawdziwą alternatywę: albo uchylimy drzwi dla cudzoziemców z naprawdę dalekich krajów - mówię głównie o Azji - którzy też są obecni w Polsce i są chwaleni jako pracownicy, albo wybierzemy dużo trudniejszą, ale chyba lepszą ścieżkę zmiany polskiego prawodawstwa w ten sposób, żeby setki tysięcy czy miliony Polaków wygnanych przez kolejne rządy z Polski za chlebem przynajmniej rozważało chęć i możliwość powrotu do Polski. Wiem, że to nie dotyczy ustawy, o której dzisiaj rozmawiamy, natomiast to są sprawy, o których powinniśmy rozmawiać przy każdej okazji.

Bardzo proszę. Pani Marszałek!

Bardzo dobrze, że ta ustawa została przygotowana.

Polska jest krajem, który w tej chwili bardzo przyciąga obcokrajowców, którzy chcą studiować na polskich uczelniach, ale również instytuty naukowe zabiegają o to, żeby można było skorzystać z doświadczeń innych naukowców. W związku z tym takie klarowne przepisy, które określają, jakie są możliwości pobytu na terenie Polski i podejmowania różnego rodzaju aktywności zawodowej, są w naszej ocenie bardzo, bardzo cenne.

Tak jak już większość moich przedmówców mówiła, ustawa nie budziła kontrowersji, w związku z tym ja tylko mogę potwierdzić fakt, że klub Nowoczesna oczywiście będzie głosować za jej przyjęciem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań posłanek i panów posłów chce wpisać się jeszcze na listę osób zadających pytania? Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! W zasadzie mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy edukacji.

I pytanie jest takie, panie ministrze: Ile jest w ciągu roku, w skali roku osób, które przyjeżdżają do Polski, uzyskują tutaj świetne wykształcenie, a następnie wyjeżdżają gdzieś indziej zarabiać pieniądze i płacą podatki w innych państwach? To po pierwsze. Proszę wybaczyć szczerość, ale ja nie jestem zwolennikiem Polski resortowej i chciałbym, żeby rząd spoglądał na problem całościowo.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Minister! Czy jednostki naukowe dysponują lub czy będą dysponowały odpowiednimi instrumentami, narzędziami, żeby móc zweryfikować prawdziwość wszelkich niezbędnych, potrzebnych informacji o cudzoziemcach, wyegzekwować je dla prawidłowego wdrożenia ww. ustawy? Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Czy w związku z proponowanymi rozwiązaniami nie ulegnie pogorszeniu bezpieczeństwo lub nie ulegną utrudnieniu działania organów monitorujących sprawy bezpieczeństwa związane z ruchem migracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem działań organów odpowiedzialnych za monitorowanie zagrożeń terrorystycznych? Temat wywołany tutaj przez kolegów, dotyczący studentów zagranicznych, studiujących w Polsce. To jest też z punktu widzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych istotne narzędzie polityki państwa polskiego, zwłaszcza w krajach afrykańskich, bo bardzo wielu studentów krajów afrykańskich studiowało przez wiele lat w Polsce. A to są osoby, które pełnią dzisiaj bardzo wysokie funkcje państwowe w krajach swojego zamieszkania. Pani poseł Zofia Czernow, Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, zada kolejne pytanie. Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Ja się cieszę, że uregulowana zostaje dosyć konkretnie sprawa cudzoziemców, którzy będą studiować, prowadzić badania naukowe w Polsce.

Szkoda, że nie udało nam się uregulować w sposób taki jak w innych krajach Unii Europejskiej kwestii określania czasu pracy cudzoziemców na podstawie uproszczonej procedury, a więc oświadczenia. Polska w tej chwili jest bardzo mało atrakcyjna w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, gdyż my mamy bardzo krótki ten czas. Resort zapowiadał wydłużenie tego okresu dla cudzoziemców, którzy ubiegają się o pracę w Polsce. Kiedy to nastąpi? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Mam kilka pytań takich technicznych. Wiemy z tej ustawy, ile będzie kosztowało Polaków, polski budżet wejście w życie tych zapisów. Natomiast nie za bardzo wiemy, co będzie kosztowało. Gdybym mógł poprosić o informacje, czy chodzi o zwiększenie zatrudnienia, czy jakieś inwestycje sprzętowe. Na co te pieniądze mają pójść? Drugie pytanie. Panie ministrze, ta ustawa ma spowodować jakby jednolitość zasad w całej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o studentów. Natomiast bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami, że obcokrajowcy, którzy są w Polsce, biznesmeni, głównie ludzie biznesu, przyjeżdżają do Polski na wizach francuskich, niemieckich, hiszpańskich, włoskich, bo twierdzą, że mimo funkcjonowania Schengen, mimo teoretycznie identycznych zasad tamtejsze wizy dostają bez problemu, natomiast polskich nie dostają, że albo mają odmowy, albo procedura trwa tak długo, że im się to nie opłaca. Dziękuję. Ostatnie pytanie w tym punkcie zada pan poseł Jerzy Meysztowicz, klub Nowoczesna. Dziękuję za możliwość zadania pytania. Większość studentów, którzy przyjeżdżają do Polski spoza Unii Europejskiej, to są osoby, które płacą za swoje studia.

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za przedłożone pytania. Pragnę na wstępie zaznaczyć, że kilka zadanych pytań tematycznie się pokrywa. Pierwsze pytanie, które zostało tutaj zgłoszone, dotyczyło obszaru projektowanej regulacji. Proszę zwrócić uwagę na to, że zasady techniki prawodawczej wprowadzone rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów wyraźnie regulują zakres tematyczny przedmiotu ustawy.

Wydaliśmy jako kraj członkowski Unii Europejskiej najwięcej zezwoleń, czyli ok. 700 tys., na pobyt ze względu na pracę - ujmuję ogólnie te dane - w związku z powyższym również ten argument nie znajduje tutaj uzasadnienia. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące liczby studentów zagranicznych, którzy obecnie podjęli studia na polskich uczelniach, w zaokrągleniu mogę podać, że jest to liczba ok. 75 tys. studentów cudzoziemskich studiujących na wszystkich uczelniach, o których mowa w Prawie o szkolnictwie wyższym, czyli chodzi o wszystkie kategorie uczelni, które ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje. Odnosząc się do pytania w zakresie bezpieczeństwa, chciałabym przywołać dyskusję, która odbyła się na posiedzeniu podkomisji komisji spraw wewnętrznych i administracji. Argumenty, które zostały przedstawione na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej, skupiały się na tym, że interes Rzeczypospolitej Polskiej każdorazowo wymaga dookreślenia w procesie stosowania danego przepisu prawa. W takim przypadku w interesie Rzeczypospolitej Polskiej może leżeć wiele wartości. Rozwój gospodarczy i dbałość o bogacenie się społeczeństwa, zapewnienie właściwego poziomu dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego musi być w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami regulującymi dbałość o dobro Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie stosunków z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Pozytywną przesłanką tego zatwierdzenia będzie skonfrontowanie stanu, w którym dany rodzaj jednostki przyjmującej będzie mógł powodować wjazd cudzoziemców w określonym celu. Będzie to konfrontacja ze stanem, w którym takie ogólne wartości są realizowane. Każda decyzja ministra spraw wewnętrznych i administracji o odmowie zatwierdzenia będzie musiała zawierać uzasadnienie i będzie podlegać kontroli w instancji odwoławczej. Mówię o instytucji zatwierdzania, która też była przedmiotem dyskusji, która odbywała się na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej. Kolejne pytanie również dotyczyło problemu cudzoziemców, czyli określania czasu pracy w formie oświadczeń.

Narzędzie wprowadzone w innej ustawie, polegające na składaniu... na podjęciu pracy na podstawie oświadczenia w Polsce jest szeroko badane i jest ono uregulowane szczegółowo również w aktach wykonawczych. Nie chcę zajmować... ponieważ jest to materia regulacji innego resortu, resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, ale na chwilę obecną, jak mówię, doprecyzowania w ustawach szczegółowych są bardzo precyzyjne.

Odnośnie do oceny skutków regulacji i zabudżetowania ustawy: są to koszty, które zostały przewidziane na obsługę cudzoziemców, są to koszty dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Kolejne zadanie. Kolejne pytanie, bardzo przepraszam, dotyczyło znikomego odsetka wydawanych wiz zagranicznych. To kwestia, która jest w obszarze polityki wizowej prowadzonej przez resort Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale pragnę. Proszę przyjąć wyjaśnienie, że jeżeli chodzi o wydawanie, podstawę wydawania wiz, tzw. wiz studenckich, jeżeli chodzi o odsetek odmów, jest on rzeczywiście znikomy.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Prawo własności przemysłowej dotyczy implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Projekt ten, druk nr 3107, 14 grudnia 2018 r. został skierowany do pierwszego czytania do Komisji Gospodarki i Rozwoju z zaleceniem przedstawienia sprawozdania. Komisja na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2019 r. rozpatrywała ww. projekt ustawy. Po przeprowadzeniu pierwszego czytania, podczas rozpatrywania ww. projektu w komisji zgłoszono szereg poprawek o charakterze legislacyjno-redakcyjnym oraz cztery poprawki o charakterze merytorycznym dotyczące art. 1 pkt 17, art. 1 pkt 22, art. 4 i art. 6, które zostały zaakceptowane przez komisję. Tak więc Komisja Gospodarki i Rozwoju rekomenduje projekt ustawy, druk nr 3121, z naniesionymi już poprawkami do drugiego czytania. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Antoni Duda, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec rządowego projektu ustawy o zmianie Prawo własności przemysłowej, druki nr 3101 oraz 3121.

Znak towarowy jest samodzielnym dobrem niematerialnym, którego istotna rola gospodarcza polega na utrwaleniu w świadomości potencjalnego odbiorcy skojarzeń wiążących nośnik oznaczenia z danym przedsiębiorstwem. W tym rozumieniu znak towarowy stanowi czynnik wpływający na innowacyjność przedsiębiorców. Potrzeba odróżnienia się od innych konkurentów prowadzi do stałego udoskonalania i rozwoju produktu. W polskim systemie prawnym zarówno przepisy prawa materialnego dotyczące znaku towarowego i prawa ochronnego na znak towarowy, jak i przepisy postępowania w sprawie dokonywania zgłoszeń i udzielania prawa ochronnego stanowią materię ustawową. Regulacje te zawarte są w ustawie Prawo własności przemysłowej. W związku z tym w celu prawidłowej implementacji dyrektywy proponuje się wprowadzenie zmian w odpowiednich przepisach tej ustawy.

Regulacja ma bardzo doniosłe znaczenie ekonomiczne i gospodarcze. W zakresie uproszczenia i zwiększenia dostępności systemu ochrony znaków towarowych nowelizacja ma objąć ok. 2 mln aktywnych przedsiębiorców i ok. 180 tys. uprawnionych z tytułu pozostających w mocy znaków towarowych. Ponadto oczekuje się, że uproszczenie sposobu przedłużania ochrony na znaki towarowe doprowadzi do zmniejszenia liczby wygaśnięć z mocy ustawy praw wyłącznych na znaki towarowe na skutek braku uiszczenia opłaty za kolejny okres ochronny. Obecnie na skutek braku uiszczenia opłaty wygasa z mocy ustawy ok. 6 tys. praw wyłącznych na znaki towarowe. Co istotne, projekt przewiduje także wprowadzenie zmian w zakresie trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Obecnie przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy wymaga złożenia pisemnego wniosku i wydania przez Urząd Patentowy decyzji. Zgodnie z proponowanymi zmianami aby przedłużyć prawo ochronne na znak towarowy, wystarczające będzie wniesienie opłaty za kolejny okres ochronny przez uprawnionego lub osobę ustawowo bądź umownie upoważnioną. Co więcej, po stronie Urzędu Patentowego wprowadzony zostaje obowiązek informowania uprawnionych z prawa ochronnego o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za kolejny okres ochronny. Ważnym skutkiem implementacji dyrektywy jest zmiana definicji znaku towarowego. Dotychczas warunek konieczny był taki, iż znakiem towarowym mogło być tylko takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, a obecnie rezygnuje się z tego wymagania. W aktualnych warunkach gospodarki i postępu technologicznego, mając na uwadze nietradycyjne znaki towarowe, np. dźwięki, znaki zapachowe czy holograficzne, taki wymóg jest przestarzały. W konsekwencji, zgodnie z nowelizowanym przepisem, znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie, jeśli będzie umożliwiało odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego i będzie możliwe przedstawienie tego znaku w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielanej na ten znak. Podsumowując, należy stwierdzić, że projektowane zmiany przyczynią się do dalszej ochrony polskich przedsiębiorców w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym, zapewniając bezpieczeństwo w obrocie znakami towarowymi. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość rekomenduję Wysokiemu Sejmowi uchwalenie ustawy o zmianie Prawo własności przemysłowej zawartej w druku nr 3121. Proszę o zabranie głosu panią poseł Aldonę Młyńczak, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! W imieniu klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska mam zaszczyt przedstawić opinię odnośnie do rządowego projektu ustawy o zmianie

Dyrektywa ma na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, a tym samym wyeliminowanie norm niezgodnych z przepisami dyrektywy.

W związku z tym transpozycja dyrektywy powinna nastąpić najpóźniej do dnia 4 stycznia 2019 r., czyli można powiedzieć, że już jesteśmy po terminie. Charakter proponowanych zmian wymaga ich ujęcia w formie przepisów ustawy z uwagi na fakt, że obejmują one prawa i obowiązki podmiotów zainteresowanych uzyskaniem ochrony lub też podmiotów uprawnionych, a także zawierają dotychczasowe regulacje w przedmiocie zgłaszania, rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, które są uregulowane w ustawie. W związku z powyższym projekt przewiduje wprowadzenie następujących zmian do systemu ochrony znaków towarowych. Przede wszystkim przewiduje rezygnację z obowiązku graficznego przedstawienia znaku towarowego, co jest związane z unowocześnieniem instytucji znaków towarowych i dopuszczeniem w ten sposób niekonwencjonalnych do tej pory znaków, jak znaki dźwiękowe, smakowe czy zapachowe. Projekt również zawiera modyfikację katalogu bezwzględnych i względnych podstaw odmowy udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe, modyfikację instytucji i zakresu ochrony znaku towarowego gwarancyjnego, a także wspólnego znaku towarowego, modyfikację zasad udzielania licencji i uprawnień licencjobiorcy, w szczególności w zakresie możliwości dochodzenia przez niego roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, czy też modyfikację roszczeń cywilnoprawnych, jakie przysługują uprawnionym z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Ponadto rozwiązania zawarte w projekcie przewidują nowe korzyści dla przedsiębiorców dotyczące w szczególności odejścia od zasady przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy na pisemny wniosek uprawnionego na rzecz uiszczania opłaty w określonym terminie. Ma to prowadzić do odformalizowania sposobu przedłużania ochrony znaku towarowego, a także do szybszego i sprawniejszego załatwiania spraw w tym zakresie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Również rozwiązania zawarte w projekcie przewidują wprowadzenie obowiązku informacyjnego Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zbliżającego się terminu uiszczenia opłaty za dalszy okres ochronny znaku towarowego. W efekcie przyjęcia nowelizacji ustawy w zakresie prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej w przedmiocie zgłaszania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych nastąpi zgodność i osiągnięty zostanie cel dyrektywy, a w szczególności dotyczący systemu ochrony znaków towarowych, który powinien być, zdaniem ustawodawców, bardziej jasny, bardziej dostępny, zrozumiały i obiektywny.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W pierwszej kolejności muszę powiedzieć, że to miłe, że akurat tylu posłów czy tyle osób, również minister z Opolszczyzny, zajmuje się tematem Prawa własności przemysłowej. Drodzy państwo, no cóż, jest to nowelizacja będąca implementacją dyrektywy, przepisów europejskich, więc tutaj zbyt dużego pola manewru nie ma, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o te propozycje przepisów, które są zawarte w tym projekcie, to one są niekontrowersyjne, dobrze kojarzone, dobrze interpretowane.

Niemniej nie byłbym uczciwy, gdybym korzystając z możliwości mówienia o Prawie własności przemysłowej, nie wspomniał o tym, że do mojego biura poselskiego zgłaszają się rzecznicy patentowi, którzy zwracają uwagę na to, że cały system ochrony własności przemysłowej nie chroni skutecznie przedsiębiorców polskich, że nie zawsze polski przedsiębiorca jest stawiany na pierwszym miejscu. Oczywiście rozumiem to, że nie jesteśmy samotną wyspą, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc funkcjonujemy w obrębie przepisów europejskich.

Z całą pewnością jeszcze do pana ministra się zwrócę w tej sprawie. Natomiast wracając do tych konkretnych przepisów - drodzy państwo, to wspominane zarówno przez przedstawiciela strony rządowej, jak i przez posłów odejście od formalności, czyli to, że znakiem towarowym nie musi być tylko znak graficzny. Może kiedyś, w dawnym ujmowaniu własności przemysłowej czy tego, co techniczne, była taka dążność, takie rozumienie, że to musi być zapisane w formie graficznej. Dzisiaj już wiemy, że nie.

Tutaj być może również warto zastanowić się nad kolejnymi nowelizacjami wykraczającymi już poza te ramy, które są nam sugerowane czy proponowane w dyrektywach, żeby w ogóle odejść od tego sformalizowania, czyli dojść do sytuacji, w której Urząd Patentowy czy urząd, który zajmuje się przydzielaniem ochrony tych praw, tak naprawdę stanie się jedynie arbitrem. I tu ostatnia kwestia, na którą zwracam uwagę z całą stanowczością.

Rzecznicy patentowi uznają za błąd sytuację, w której sądy powszechne, które są powoływane do sądzenia w zasadzie we wszystkich sprawach. Jednak jest dosyć duża specyfika spraw z zakresu Prawa własności przemysłowej. A więc przekazuję zapytanie, kiedy faktycznie takie sądy zaczną w sprawny sposób funkcjonować w Polsce, tak żeby własność przemysłowa, czyli tak naprawdę prawa i interesy polskich przedsiębiorców, była chroniona w sposób należyty, przez sądy i sędziów, którzy będą wyspecjalizowani stricte w tym konkretnym kierunku, po to aby w jak najpełniejszy sposób chronić interes polskich przedsiębiorców, polskich wynalazców, polskich producentów, wszystkich tych, którzy pracą swojego umysłu, swoich mięśni, maszyn, które konstruują i z których korzystają, budują tak naprawdę bogactwo naszej ojczyzny. Proszę o zabranie głosu pana posła Jerzego Meysztowicza, klub Nowoczesna. Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić opinię klubu Nowoczesna co do druku nr 3107, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej. Prawo własności przemysłowej wynika z konieczności implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. To bardzo ważne, że w tej chwili ministerstwo, Urząd Patentowy podjęły się przygotowania tej ustawy, ponieważ ona nie tylko doprowadza do sytuacji, kiedy te prawa zostają ujednolicone, ale również zmienia się sytuacja, jeśli chodzi w ogóle o ochronę wartości przemysłowej, dlatego że zmieniają się techniki, zmienia się technologia, zmieniają się różne formy, również różne formy znaków towarowych.

Chciałbym podkreślić tutaj bardzo dobrą współpracę między ministerstwem i Urzędem Patentowym. Także na posiedzeniu komisji mieliśmy okazję wysłuchać kilku uwag ze strony rzeczników patentowych. Jedna z ich poprawek została nawet uwzględniona. To świadczy o tym, że ta ustawa została dobrze przygotowana i we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi. Uważam, że to jest cenne działanie, aby polska myśl techniczna, polskie firmy, polskie towary były chronione, żeby nie tylko wiedzieć, na jakich zasadach można ubiegać się o ochronę ze strony polskiego prawa, ale również wiedzieć, że na tych samych zasadach można ubiegać się o ochronę także ze strony praw europejskich. Ciekawe jest to, że odchodzi się od takich rzeczy jak konieczność przedstawiania znaku towarowego w formie graficznej. Dobrze, że zostały określone warunki wykorzystania wspólnego znaku towarowego. Te wszystkie zmiany, wydaje się, służą temu, aby polska myśl techniczna, polski przemysł i polscy przedsiębiorcy mieli sposobność ochrony swojej własności intelektualnej. Czy ktoś z państwa chciałby się jeszcze dopisać na liście osób zadających pytania? Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Paweł Grabowski, klub Kukiz’15.

Wysoka Izbo! Moje pytanie będzie dotyczyło właśnie sądownictwa z zakresu prawa własności przemysłowej: Jakie konkretnie są pomysły, jeżeli takie są? A jeżeli ich nie ma, to kiedy możemy się spodziewać podjęcia tego tematu przez ministerstwo czy też przez rząd? Ponieważ, tak jak mówię, rzecznicy patentowi zwracają uwagę na to, że często niestety nie ma odpowiedniego poziomu zrozumienia dla skomplikowania albo bardziej specyfiki, właściwie nie dla skomplikowania, ale specyfiki spraw z zakresu prawa własności przemysłowej.

Pytanie zadaje teraz pan poseł Jarosław Gonciarz, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Pytanie: Jak zmiany w procedowanym projekcie ustawy Prawo własności przemysłowej wpłyną na pozycję polskich przedsiębiorstw? Czy będą miały wpływ na tendencję ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki europejskie, czy będą miały wpływ na rozpoznawalność polskiej marki na arenie europejskiej? Pytanie zadaje pan poseł Piotr Pyzik, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać o ewentualne sprawy sporne. Jak przedłożony projekt wpłynie na rozwiązywanie ewentualnych spraw spornych w przypadku złożenia przez Urząd Patentowy sprzeciwu wobec wyznaczenia na terytorium Polski międzynarodowego znaku towarowego? A jak w przypadku odwrotnym, kiedy odpowiedni urząd innego państwa Unii Europejskiej wniesie taki sprzeciw wobec wniosku polskiego przedsiębiorcy? Pytanie zadaje pani poseł Zofia Czernow, PO-KO. Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Chciałam zapytać o statystykę, kilka krótkich pytań. Pierwsze pytanie: Ile w minionym roku wpłynęło zgłoszeń o ochronę znaku towarowego? Drugie: Jaka to jest dynamika w ostatnich 5 latach? Trzecie pytanie: Ile wpłynęło zgłoszeń dotyczących rejestracji ochrony znaku międzynarodowego? I ostatnie pytanie: Jaki jest średni czas oczekiwania na wydanie decyzji zwłaszcza w przypadku pierwszego wniosku, o nową rejestrację? Pytanie zadaje pan poseł Paweł Skutecki, klub Kukiz’15. Panie Ministrze! Tylko w związku z tym muszę zadać jedno pytanie: w tej ustawie jest zapisane, że wchodzi ona w życie 1 dzień po opublikowaniu. Nie ma żadnych obaw co do przedsiębiorców, bo oni na pewno będą gotowi, ale czy zdaniem pana ministra Urząd Patentowy też będzie gotowy?

Szanowna Panie Marszałek! Bardzo dziękuję za wszystkie głosy w dyskusji i wszystkie pytania.

Ja mogę powiedzieć, że ten temat jest przedmiotem prac specjalnego zespołu, dlatego że ten postulat znalazł się w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, więc my tak samo zidentyfikowaliśmy ten problem i - nie chciałbym się wypowiadać w imieniu gospodarza tego tematu - mogę tylko powiedzieć, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii aktywnie uczestniczy w pracach tego zespołu i popiera postulat utworzenia sądów do spraw własności intelektualnej jako tych, które będą w sposób profesjonalny szczególnie przyglądać się sprawom, których dotyczy także przedmiot tej ustawy. Oczywiście wpływy tej ustawy są niebagatelne, dlatego że regulacja w zakresie upraszczania i zwiększania dostępności systemu ochrony znaków towarowych, co sami państwo posłowie podnosiliście, ma objąć swoim zakresem ok. 2 mln aktywnych przedsiębiorców i 180 tys. uprawnionych z tytułu pozostających w mocy znaków towarowych. Tak więc zakres jest bardzo szeroki i z pewnością przedsiębiorcy czekają na te regulacje. Stąd nie ma kontrowersji wokół tej ustawy i ona cieszy się poparciem, dlatego że wszyscy na nią czekali.

Jeśli chodzi o wejście w życie ustawy, to w związku z tym, że te regulacje są oczekiwane przez przedsiębiorców, jesteśmy za tym, żeby czas wejścia w życie był jak najkrótszy, dlatego że ustawa poszerza wolności obywatelskie, sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej, jest po prostu wyczekiwana przez przedsiębiorców i stronę społeczną.

Szanowni Państwo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych chciałem złożyć sprawozdanie z prac nad ustawą o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Dokonaliśmy znaczącego przeglądu przepisów dotyczących dyrektyw unijnych, dlatego że jest to kolejna ustawa, która jest formą implementacji dyrektywy unijnej.

W związku z tym należy obecnie, przystępując do końcowej fazy prac, zgłosić pewne zmiany do tej ustawy. One zostaną przedłożone w formie poprawek klubu parlamentarnego. Ponieważ będę występował również w imieniu klubu, nie chciałbym zabierać więcej czasu. Ustosunkuję się do tych zmian i samego projektu zmiany ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w wystąpieniu klubowym. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwszy pan poseł Jan Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! To kolejna duża próba legislacyjna, duży projekt legislacyjny wynikający z naszych zobowiązań implementacyjnych dotyczących dyrektyw unijnych.

Ten projekt ma na celu usprawnienie już wprowadzonych rozwiązań związanych z procesami restrukturyzacyjnymi. Wprowadza również pewne znaczące uściślenia, uregulowania, doprecyzowania w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Dotyczy to także kwestii uprawnień w ramach restrukturyzacji banku zrzeszającego, kwestii utworzenia instytucji pomostowej i funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów, jak również możliwości krzyżowego wykorzystywania funduszy gwarancyjnych banków i kas oszczędnościowo-kredytowych.

To niezwykle skomplikowane procedury sanacyjne i restrukturyzacyjne. One wprowadzają dodatkową kategorię wierzytelności z tytułu długu nieuprzywilejowanego w ramach postępowania upadłościowego w celu usprawnienia procesu przymusowej restrukturyzacji, w szczególności w aspekcie ewentualnego procesu umarzania lub konwersji tego typu zobowiązań.

Z uwagi na nieprowadzenie przez nie tej działalności depozytowej, w przypadku upadłości banku hipotecznego nie będzie występował przypadek wypłaty środków gwarantowanych. Doprecyzowano cały szereg definicji.

Uzupełnia się katalog definicji stosowanych w ustawie o BFG w zakresie zobowiązań zabezpieczonych.

Wprowadza się możliwość przyjęcia grupowego planu przymusowej restrukturyzacji w ramach tzw. wspólnej decyzji w sytuacji, gdy podmiotem zależnym jest właśnie podmiot będący podmiotem znaczącym.

Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią poseł Izabelę Leszczynę, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! To miał być zwyczajny projekt wdrażający dyrektywę unijną, projekt, który wprowadza przepisy ułatwiające stosowanie procedury resolution, czyli procedury przymusowej restrukturyzacji w bankach zagrożonych upadłością czy bankach, które nie są wystarczającym gwarantem bezpieczeństwa depozytów swoich klientów.

Co więcej, zrobiliście to w dwóch ustawach na raz.

Były dwie zupełnie odrębne ustawy. Jedna dotyczyła Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i procedury resolution, druga - nadzoru nad rynkiem finansowym. Typowy plan Zdzisława z taśm, których nie zdołało zagłuszyć szumidło pana Chrzanowskiego. Okazało się, że tamta wyszła pierwsza. Zrobiło się wam wstyd.

Nikogo nie interesuje to, co dzisiaj dzieje się w polskim Sejmie, więc doszliście do wniosku, że to jest najlepszy moment, żeby cichaczem przemknąć z tą ustawą wstydu. żeby już o tym planie Zdzisława nie mówić. Ale mylicie się. Wy zostaniecie z tym wstydem, a my będziemy wam patrzeć na ręce. Będziemy wam patrzeć na ręce zarówno wtedy, gdy będziecie sprzedawać jakiś bank za złotówkę, jak również będziemy wam patrzeć na ręce, gdy będziecie sprzedawać SKOK Wołomin za złotówkę. Będziemy patrzeć wam na ręce, jak będziecie ukrywać listy kredytobiorców SKOK-u Wołomin. Będziemy patrzeć wam na ręce wtedy, gdy sprzedając SKOK Wołomin, pozbawicie BFG możliwości odzyskania pieniędzy wypłaconych na gwarancje. Będziemy patrzeć na ręce zarówno panu Sokalowi w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, jak i następcy pana Chrzanowskiego.

Co się dzieje dalej z propozycją korupcyjną, którą złożył pan Marek Chrzanowski? Dlaczego właściwie w ustawie budżetowej dzisiaj, co nie zdarzyło się nigdy, KNF dostaje dotację podmiotową w wysokości 75 mln? I dlaczego polski podatnik ma za to płacić?

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kilka słów opinii co do sprawozdania komisji o tym rządowym projekcie.

Wyłączenie banków hipotecznych z systemu gwarancyjnego, bo i po co, jeśli nie ma tam depozytów, wprowadził między innymi, usprawnił restrukturyzację banku zrzeszającego poprzez stworzenie instytucji pomostowej, ochroną gwarancyjną objął również rachunki bankowe rad rodziców przy szkołach. Ale w tej zasadniczej, podstawowej wersji projektu, powiem szczerze, nie staraliśmy się doszukiwać jakichś ukrytych zmian, które niekoniecznie mają za zadanie implementację, interpretację czy usprawnienie procesów gwarancyjnych w systemie bankowym. A zgłoszone do projektu poprawki niestety budzą bardzo wiele uwag i kontrowersji, tym bardziej że niedawno przyjęta ustawa pod bardzo ładnym tytułem: „wzmocnienie nadzoru oraz ochrona inwestorów na rynku finansowym”, miała na celu bynajmniej nie ochronę inwestorów, ale likwidację przez Komisję Nadzoru Finansowego instytucji bankowych według niedopuszczalnych w naszej ocenie zasad korupcyjnych wzmacnianych urządzeniem zwanym szumidłem.

Na taśmach z KNF-u mówi się o pomysłach, projektach Zdzicha. I pytanie jest jasne: Czy to jest tylko zbieg okoliczności, czy swoimi działaniami chcecie przykryć aferę kilku instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo finansowe Polaków, bo tak naprawdę dzisiaj chyba tylko naiwni mogą uwierzyć, że afera KNF-u dotyczy wyłącznie pana Chrzanowskiego? Omawiany dzisiaj projekt gwarantuje środki na wzmocnienie finansowe nie banków restrukturyzowanych, wymagających takiego wsparcia, nawet banków podlegających tzw. przymusowej restrukturyzacji, co jest oczywiste, ale banków przejmujących te inne. Jak się okazuje, przejmujących je za złotówkę. Projekt ułatwia także swobodne korzystanie ze środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez upadające SKOK-i, a ze składu Zarządu BFG wyeliminowano już przedstawicieli Związku Banków Polskich, a więc tych jednostek, które tworzą Bankowy Fundusz Gwarancyjny, i oczywiste wydaje się, że ich obecność w BFG jest uzasadniona. W ogóle nasuwa się pytanie, dlaczego dotychczas przy tych różnych patologiach w systemie SKOK-ów nie ma wciąż komisji śledczej. To przecież SKOK-i dotyka niewypłacalność i upadłość. Przypomnę, że opłaty SKOK-ów na rzecz BFG utrzymane są nadal na kilkakrotnie niższym poziomie niż opłaty np. małych, polskich banków spółdzielczych, a ten projekt zakłada dalsze preferencje właśnie dla SKOK-ów. Tego projektu nie można rozpatrywać odrębnie, w oderwaniu od przyjętych już uregulowań dotyczących zarówno BFG, jak i Komisji Nadzoru Finansowego. Tutaj pod przykrywką złudnych haseł destabilizuje się finanse państwa, wprowadza niepokój, urzeczywistnia cele, które są wyłącznie realizacją nieujawnionych, nikczemnych strategii wymyślonych przez rządzących. Jesteśmy przekonani, że projekt analizowanej ustawy nie jest niewinnym aktem prawnym, który cokolwiek dobrego chce wprowadzić czy usprawnić w systemie [[Dzwonek]] gwarancji bankowych. Proszę o zabranie głosu panią poseł Paulinę Hennig-Kloskę, klub Nowoczesna.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Dwa miesiące zajęło wam wprowadzenie z powrotem tego projektu pod obrady, bo szukaliście takiego tygodnia, w którym cała opinia publiczna w Polsce będzie zajęta czymkolwiek innym, a nie tym, co dzieje się w Sejmie. Niestety tragiczne wydarzenie ostatnich dni wy wykorzystujecie do tego, aby pchać przez ten Sejm kolejny niewygodny, bardzo niewygodny dla was, temat, czyli kwestię tej słynnej poprawki, już dzisiaj wprowadzonej do polskiego prawa, która umożliwia sprzedaż w Polsce banku za złotówkę, czyli realizację planu Sokala. Wstyd, że wykorzystujecie tragedię, którą przeżywają dzisiaj Polacy, do realizacji takich właśnie. planów. To prawda, że ta ustawa miała być zwykłą ustawą wdrażającą poprawki do dyrektywy resolution, która ma nam pomóc wychodzić z trudnych momentów na rynku finansowym, natomiast to też prawda, że wyście jak zawsze wepchnęli do niej coś, co niezgodnie z dyrektywą tak naprawdę wprowadzało szybką ścieżkę uwłaszczania polskich banków, bo tak to trzeba nazwać. Przypomnijmy, co było w tej poprawce. Ona daje możliwość, na wypadek obniżenia sumy funduszy własnych banków poniżej wymogów kapitałowych albo powstania niebezpieczeństwa takiego obniżenia się tej sumy - bardzo niedoprecyzowane pojęcie - Komisji Nadzoru Finansowego podjęcia decyzji o przejęciu banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego. Przypomnijmy Polakom, jak to było. Nie jest realizacja dyrektywy, bo kwestie dotyczące przejmowania, restrukturyzacji, a potem kontrolowanego przejmowania banków będących w trudnej sytuacji finansowej już w polskich przepisach mamy. Nie dotyczy to małych banków spółdzielczych, jak przez chwilę posłowie Prawa i Sprawiedliwości próbowali wmawiać opinii publicznej, to jest po prostu realizacja planu Sokala. Ktoś wdusił Ministerstwu Finansów pod hasłem realizacji dyrektywy przepisy, na których najwyraźniej zależało panu Chrzanowskiemu, bo przypomnijmy, że to on osobiście zabiegał o to, aby te poprawki pilnie znalazły się najlepiej w pięciu ustawach, bo która pierwsza zostanie przyjęta, ta lepsza. Nie udało się. Słynne taśmy, których nie zagłuszyły szumidła pana Chrzanowskiego, usłyszała opinia publiczna i zaczął się młyn. Ustawa co posiedzenie miała znaleźć się w harmonogramie naszych obrad, ale co posiedzenie znikała, nie było takiej okazji jak dziś. Dzisiaj złożę poprawkę, która będzie z polskiego prawa usuwała szybką ścieżkę uwłaszczania banków. Będziemy to piętnować przy każdej okazji. Nie ma zgody na sprzedawanie SKOK-u Wołomin na złotówkę. Co najlepsze, szanowni państwo, w trakcie tego całego zamieszania w KNF, właśnie wtedy, kiedy w KNF panowało bezkrólewie, pełniący raptem 8 dni obowiązki szefa KNF pan Marcin Pachucki podjął decyzję, wydał zgodę na sprzedaż SKOK-u Wołomin za złotówkę, co sugeruje opinii publicznej i potencjalnym nabywcom, że tam nic nie ma, w zasadzie więcej długów niż majątku. Natomiast nie jest tak, bo ta oferta nie obejmuje zobowiązań wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co istotnie zmienia wycenę. Chcecie sprzedać 3 mld kredytów za 92 mln, 1 mld hipotek, co nagle zostało wycenione przez nikomu nieznaną spółkę, mimo że cały operat szacunkowy SKOK-u Wołomin robił Uniwersytet Szczeciński, nagle ten dziwnie wyceniony portfel hipotek... 1600 hipotek chcecie sprzedać za 72 mln. Nawet odejmując hipoteki wyprzedzające, panie ministrze, tam zostaje 600 mln czystej hipoteki do sprzedaży. Nie wiem, kto to wyceniał i w oparciu o jakie metody, ale sprawdzimy to, bo Komisja Finansów Publicznych zajmie się tym w lutym. Składam również dwie poprawki. Uważam, że w związku z tymi ostatnimi wydarzeniami w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powinni znaleźć się [[Dzwonek]] przedstawiciele Związku Banków Polskich. Przechodzimy do zadawania pytań.

Chciałam zadać dwa pytania dotyczące najbardziej kontrowersyjnych zapisów w tym projekcie. Pierwsze pytanie dotyczy tego, co dalej z zapisem wprowadzonym do projektu ustawy, który pozwala przejmować bank w trudnej sytuacji, zagrożony upadłością, za złotówkę.

Druga poprawka.

Wysoka Izbo!

Otóż na początku wszystkie banki, które wpłacały składki do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, mogły zaliczyć te składki do kosztów uzyskania przychodów, później państwo to zmieniliście. Chciałem się dowiedzieć dlaczego państwo uważacie, że to jest niesprawiedliwe i że banki nie mogą odliczać tego z kosztów uzyskania przychodu. Mam nadzieję, że państwo uwzględnicie poprawkę zgłoszoną przez moją koleżankę z klubu Nowoczesna i przywrócicie możliwość odliczania tej składki od podstawy i od kwot dochodu. Jako kolejny pytanie zada pan poseł Mirosław Suchoń, klub Nowoczesna. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Trudno uciec od takiego wrażenia, że jednak powrócenie tej ustawy nie jest przypadkiem. Muszę powiedzieć, że czuję się bardzo zbulwersowany, ponieważ przy okazji. Pan wie o tym, że wszystko było uzgadniane i nikt nie zgłaszał sprzeciwu co do takiego procedowania. Bardzo proszę. Pani Marszałek!

Jednak warto, panie ministrze, aby przedstawiciel resortu jeszcze raz stanął przed nami i przedstawił swoje stanowisko dotyczące wyceny majątku SKOK-u Wołomin, zaproponowanej ceny wywoławczej [[Dzwonek]] za sprzedaż tego SKOK-u, bo to jest sprawa, która absolutnie bulwersuje opinię publiczną.

Szanowni Państwo!

Komisja Europejska, która sprawdzała, czy mamy to wszystko zaimplementowane, tak jak powinno to być zrobione, uznała, że pewne rzeczy trzeba poprawić.

Środowiska bankowe - a państwo tak to tutaj przedstawiacie, że bank może być przejęty za złotówkę - popierają ten przepis, czyli podmioty, których dotyczy ten przepis mówią: To jest bardzo dobry przepis.

Jeśli jest jakiś podmiot, który ma problem, KNF wysyła informację do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który pełni funkcję resolution, jest to organ resolution, i on sprawdza, czy jest w tym interes publiczny czy nie. Jeśli podmiot jest mały, zwykle tam nie ma interesu publicznego, jest upadłość.

I wtedy rozwiązaniem jest upadłość i nie ma ścieżki powrotu.

Tak więc tutaj mamy kompletny rozdźwięk. Padał zarzut, że Związek Banków Polskich nie uczestniczy w pracach Rady BFG.

Natomiast od 2016 r. z powodu implementacji dyrektywy jest to również organ resolution, który podejmuje kluczowe decyzje dotyczące właśnie przejmowania banków czy uporządkowanej likwidacji. Tak więc żeby być w zgodzie z instytucjami międzynarodowymi, czyli Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Bankiem Światowym, bo oni prowadzą tę misję..., zaimplementowaliśmy ich zalecenia. Byłoby to kompletnie nielogiczne. Stanowi to implementację zaleceń, najwyższych standardów, jeśli chodzi o stabilność sektora finansowego i sieci bezpieczeństwa. Tu zupełnie nie rozumiem tych protestów. Jeśli chodzi o przejmowanie czy. Proszę państwa, to jest plan Komisji Europejskiej, ponieważ implementacja dyrektywy właśnie mówiąca o uporządkowanej likwidacji czy przejmowaniu banków, nieważne czy to. Proszę zauważyć, że Banco Popular w Hiszpanii został przejęty przez Santander za 1 euro. Więc jeśli państwo nie zgadzacie się z tym, z tego typu dyrektywami, protestujcie w Brukseli.

Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druki nr 2770 i 3074) Proszę panią poseł Ewę Szymańską o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych, druk nr 2770. Komisja do Spraw Petycji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu skierowała do marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych. Projekt ten powstał w Komisji do Spraw Petycji w odpowiedzi na otrzymaną od Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego petycję skierowaną do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącą przeznaczenia większej niż do tej pory środków publicznych na wsparcie rozwoju turystyki w Polsce. Marszałek Sejmu zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował w dniu 18 lipca 2018 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych do pierwszego czytania. Komisja Finansów Publicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 21 listopada oraz 5 grudnia 2018 r. wnosi, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić załączony projekt ustawy. Dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Jarosław Krajewski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić nasze stanowisko w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych. Projekt ustawy, tak jak wspominała pani sprawozdawca komisji, jest reakcją na petycję skierowaną do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zgodnie z art. 63 konstytucji, o czym warto przypomnieć również w tym momencie, każdy ma prawo składać petycje w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej. I tak stało się w tym przypadku. Tu mamy do czynienia z takim solidnym przykładem, kiedy Sejm, a dokładnie Komisja do Spraw Petycji zgłosiła inicjatywę ustawodawczą, która - jak myślę - jest takim potwierdzeniem, że obywatele również mają możliwość partycypacji w procesie stanowienia prawa. Ten projekt ustawy ma zwiększyć wydatkowane środki publiczne na wsparcie rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki społecznej. Myślę, że bardzo cennym elementem tej ustawy jest kwestia zwiększenia, nawet niewielkimi nakładami finansowymi, możliwości wsparcia dostępności turystyki społecznej, rozpropagowania form aktywnego wypoczynku nieopodal miejsca zamieszkania czy ma to też poprawić infrastrukturę tysięcy kilometrów szlaków turystycznych. To jest przede wszystkim propozycja rozszerzenia katalogu podmiotów i zwiększenia liczby beneficjentów, jeśli chodzi o Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, o te wydatki, które będą przeznaczane dla podmiotów, które będą działały zgodnie z zasadą turystyki społecznej, czyli tej, która jest bez barier infrastrukturalnych, jak również pozbawiona jest barier finansowych. Jeśli spojrzymy na kwestie związane z potrzebą wspierania aktywności turystycznej, jeśli chodzi o szczególne uwzględnienie osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, to warto również spojrzeć na dane, które wskazują, że część polskich rodzin nadal nie jest w stanie sfinansować pobytu swoich dzieci, jeśli chodzi o taki w pełni komercyjny wypoczynek. Ta oferta i to rozwiązanie, które - jestem przekonany - zostanie przyjęte przez Wysoką Izbę, ma zmierzać właśnie do tego, żeby liczba podmiotów, która będzie mogła skorzystać z tego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wzrosła. Jeżeli spojrzymy na ostatnie lata, to w ramach części 40. budżetu państwa: Turystyka te wydatki były utrzymane na poziomie ok. 50 mln zł. Z tego jedynie ok. 2,5 mln zł zostało przeznaczone na bezpośrednie dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki. Omawiany projekt ustawy ma spowodować rozszerzenie tego katalogu celów o wydatki wspierające rozwój turystyki społecznej. W opinii naszego klubu jest to krok w dobrym kierunku, który w tej nieodległej przyszłości również spowoduje takie widoczne wsparcie turystyki społecznej.

Ważne jest to, że z tych środków będą mogły skorzystać zarówno samorządy, jak i organizacje pozarządowe. Myślę, że to jest to bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli dodamy do tego ten pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw, związany ze zwiększaniem aktywności turystycznej i aktywności fizycznej, to myślę, że wszystkie kluby parlamentarne poprą ten projekt ustawy.

Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić opinię klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska co do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych, druki nr 2770 i 3074.

Tak jak mój przedmówca wyrażam swoje wielkie zadowolenie z tego powodu, że można uczestniczyć w procesie legislacyjnym również w ten sposób. Muszę powiedzieć, że w pierwszej chwili, kiedy dowiedziałam się o tym projekcie, byłam bardzo mocno sceptyczna.

Bardzo wiele dzięki tym środkom udało się w Polsce zrobić. Natomiast po przemyśleniu uznałam, że rzeczywiście jest tak, że stan infrastruktury turystycznej jest nadal niezadowalający, nadal mamy bardzo wiele do zrobienia. W związku z tym otworzenie FRKF-u również na możliwość budowy, remontów i modernizacji infrastruktury turystycznej jest dobrym pomysłem. Wspomnę, że podczas właściwie wszystkich posiedzeń komisji kultury fizycznej i sportu, w których uczestniczyłam, wszystkich tych posiedzeń, na których rozpatrywane były proponowane budżety, pojawiały się wnioski o zwiększenie środków na turystykę, zwiększenie środków właśnie na infrastrukturę turystyczną.

Szlaki rowerowe górskie, dostęp do akwenów wodnych, stanice kajakowe, dostosowanie infrastruktury turystycznej do osób z niepełnosprawnościami - to jest bardzo duże, bardzo ważne zadanie, które przez nami stoi. Ministerstwo Sportu i Turystyki, pan minister zobowiązał się do tego, żeby duża część tych środków była rzeczywiście przeznaczana na infrastrukturę turystyczną. Uważam, że ono jest ważne.

Mamy nadzieję, że rzeczywiście dzięki tej ustawie, dzięki wspólnym naszym wysiłkom uda się poprawić infrastrukturę turystyczną. W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej chciałabym zadeklarować, że mój klub będzie popierał tę ustawę.

Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Nowoczesna w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych, druki nr 2770 oraz 3074. Wysoka Izbo! Przedmiotowy projekt ustawy rozszerza katalog celów, na jakie mogą być przeznaczone środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o wydatki wspierające rozwój turystyki społecznej. Ustawa, projekt ustawy został przedstawiony przez komisję na podstawie wniosku skierowanego przez PTTK.

Wysoka Izbo! W ramach projektowanej ustawy pojawi się również zapis o tym, że warunki uzyskiwania dofinansowania będą ustalane przez właściwych ministrów oraz - to już z uzasadnienia - dojdzie do zmiany rozporządzenia uwzględniającej te nowe zadania.

Oczywiście to są bardzo ważne zadania.

Jak wiemy, w górach wiele nie trzeba, ale jednak schroniska czy miejsca noclegowe, oznaczenia szlaków są elementem niezbędnym i w naszej tradycji korzystanie z tej infrastruktury jest absolutnie ważne.

Jak wiemy, decyzje w sprawach dofinansowania w roku wyborczym mogą być obarczone pokusą, powiedziałbym, sfinansowania tych zadań tam, gdzie jest to potrzebne z punktu widzenia interesów jednej czy drugiej formacji politycznej. Pragnę zaapelować w imieniu ludzi gór, miłośników gór, miłośników przyrody o to, aby ministerstwa unikały nacechowania decyzji właśnie takimi przesłankami, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi potrzebami.

Jako pierwsza pytanie zadaje pani poseł Zofia Czernow, PO-KO. Panie Ministrze! Mieszkam w Karkonoszach i bardzo często jestem w górach.

To jest absolutnie widoczne gołym okiem i jest tak od lat.

Chciałabym zapytać, kiedy będzie wiadomo, jaka kwota w ramach tegorocznego funduszu zostanie przeznaczona na turystykę społeczną. Pytanie zadaje pani poseł Joanna Mucha, PO-KO.

Drugie pytanie: Jak to procentowo będzie się układało, czyli jaka część FRKF pana zdaniem powinna zostać przeznaczona na turystykę?

Pytanie zadaje pan poseł Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek!

Chcę także zapytać o to, czy środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będą mogły być przeznaczone w ramach wsparcia turystyki społecznej na infrastrukturę turystyczną i w jaki sposób.

Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pan poseł Jerzy Meysztowicz, klub Nowoczesna. Wysoka Izbo!

Drugie pytanie: Dlaczego państwo nie zdążyliście z przeprowadzeniem tej ustawy przez Sejm?

Proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki pana Jana Widerę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rozpocznę od odpowiedzi na pytanie ostatnie: Czy środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach turystyki społecznej będą mogły być przeznaczane na infrastrukturę turystyczną? Tak, zaproponowane brzmienie art. 86 ust. 4 ustawy o grach hazardowych w wersji zaakceptowanej przez komisję to umożliwia. Jeżeli chodzi o konkretyzację zadań, będzie ona corocznie, w zależności od aktualnych potrzeb, ustalana w programie dotacyjnym ministra. Nie można zatem wykluczyć dofinansowania zadań dotyczących realizacji infrastruktury turystycznej. Konkretyzacja zadań oraz ich zasięg będą też zależały od ustalonej w programie puli środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na dofinansowanie turystyki społecznej. Odpowiadając na pytania pozostałych państwa posłów - one skumulowały się tutaj w jedną moją odpowiedź - chciałem powiedzieć, że szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, czyli tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, uwzględniają racjonalność i ciągłość finansowania zadań oraz kontroli sposobu wydatkowania ze środków funduszy. A więc wszystko to będzie określone w rozporządzeniu ministra i będzie konsekwencją konsultacji publicznych z PTTK-ami i innymi zainteresowanymi interesariuszami.

Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą. Proszę o zabranie głosu pana posła Roberta Majkę, niezrzeszonego.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Serdecznie witam obecnych na galerii naszych piłsudczyków z Ciechanowa. Szanowni Państwo! Do Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej należy ok. 5 tys. osób działających w kraju i za granicą. Jego celem jest m.in. propagowanie czynu i myśli Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, jak też wychowanie młodzieży.

Doceniam rolę edukacyjną, jaką członkowie tego stowarzyszenia pełnią w życiu społecznym. Ich obecność na uroczystościach państwowych, rocznicowych i świętach kościelnych wzbudza zainteresowanie, co ważne, u młodego pokolenia. Charakterystyczne szare mundury, maciejówki i towarzysząca temu słynna pieśń Legionów „My, Pierwsza Brygada” wzbudzają podziw, szacunek i uczucia patriotyczne. Piłsudczycy zapraszani są chętnie do szkół, gdzie uczą młodzież historii powstania Niepodległej. Kultywując pamięć marszałka Józefa Piłsudskiego, przekazują wartości tak ważne dla każdego Polaka: miłość i oddanie dla Polski. Miałam zaszczyt uczestniczyć w IV Pielgrzymce Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę w sierpniu ub.r. W roku 2018 pielgrzymowanie miało szczególne znaczenie: obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 30-lecia Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. W dowód uznania i szacunku dla zaangażowania w kultywowanie pamięci o marszałku i jego żołnierzach, przekazywanie młodzieży wzorców patriotyzmu, ofiarności i umiłowania ojczyzny ufundowałam i przekazałam w trakcie uroczystości kompletny mundur piłsudczyka ciechanowskiemu oddziałowi związku. Szczytna idea, zapał i zaangażowanie członków związku już przynoszą owoce. Coraz więcej jest młodych twarzy w szarych mundurach - godnych następców żołnierzy marszałka.

Wysoki Sejmie! Śmierć pana prezydenta Pawła Adamowicza była dla nas szokiem i druzgocącą informacją. Ja do tej pory nie mogę się z tym pogodzić.

Prezydent Adamowicz był człowiekiem szanowanym, który zawsze kierował się tolerancją, otwartością i szacunkiem dla drugiego człowieka - nawet w trudnych momentach politycznych sporów, co w Polsce jest rzadkością. Paweł Adamowicz swoją drogę naprawdę wielkiego samorządowca zaczynał w 1990 r. w Radzie Miasta Gdańska. W następnej kadencji rady został jej przewodniczącym.

Odbyliśmy też wiele inspirujących rozmów na temat rozwoju Gdańska, za co jestem wdzięczna i co zostanie we mnie na zawsze. W kolejnej kadencji Paweł Adamowicz został prezydentem miasta, które ukochał bardzo, czyli naszego Gdańska, i był nim z sukcesem przez ponad 20 lat. Panie Prezydencie! Chcę ci tą drogą, publicznie w Sejmie podziękować za 25 lat współpracy. Wiele się od ciebie nauczyłam.

W dniu 22 czerwca 2017 r. uchwalona została przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Przez pomniki zgodnie z ustawą rozumie się również kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty, tablice pamiątkowe, napisy i znaki.

Cieszyliśmy się, że po wielu latach zabiegów, starań i działań środowisk patriotycznych dokonała się sprawiedliwość dziejowa, ale już wtedy miejscy urzędnicy zapowiadali, że ten pomnik wróci. Wybory samorządowe sprawiły, że w magistracie nic się nie zmieniło i pierwszą rzeczą, która została zrealizowana tuż przed świętami Bożego Narodzenia, było wystawienie pomnika na widok publiczny. Przed ogrodzeniem radzieckiego cmentarza wojennego, przy jednej z głównych ulic miasta - ul. Wrocławskiej wybudowano betonowy podest, na którym umieszczono pomnik. Na specjalnych podstawach umocowano tablice, które wcześniej były jego na cokole. Postawiono uprzątnięte wcześniej z innych miejsc obeliski poświęcone zbrodniczym formacjom komunistycznym.

Tym sposobem pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej wrócił do przestrzeni publicznej. Przecież zawsze można powiedzieć, że został wystawiony na widok publiczny w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej, naukowej lub o podobnym charakterze w celu innym niż propagowanie ustroju totalitarnego. Przecież jest to zgodne z ustawą. Mam nadzieję, że zarówno wojewoda dolnośląski, jak i Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zainteresują się tym haniebnym legnickim pomnikiem, właściwie zinterpretują przepisy ustawy i zniknie on z przestrzeni publicznej na zawsze.